Wysoka Izbo! Wniosek formalny o stwierdzenie kworum. Wczoraj prosiliśmy panią marszałek, żebyśmy zajęli się tym, co najbardziej istotne, właśnie w obawie o to, że parlamentarzyści nie będą w stanie w sposób zdalny dobrze pracować nad tym projektem ustawy. Dlatego chciałbym od pani marszałek uzyskać informację, w jaki sposób pani marszałek jest w stanie stwierdzać to, czy obrady są zgodne z prawem, tzn. czy udział w nich bierze wystarczająca liczba posłów, czy jesteśmy w stanie na każdym etapie potwierdzić, że jest nas więcej aniżeli połowa. To raz. Gdyby pani marszałek zechciała pokazać, udowodnić, że w tej chwili każdy z parlamentarzystów może pracować. Wczoraj zgłaszaliśmy wiele uwag do systemu informatycznego, m.in. mówiąc o tym, że są problemy z udostępnianiem transmisji Sejmu, m.in. uwagi do tego, że jednoczesne zalogowanie w systemie do głosowania powoduje zerwanie transmisji obrad, czyli że poseł de facto jest bez informacji. W tej chwili posłowie sygnalizują, że sygnał, który mają, jest z opóźnieniem, więc to, co dzieje się na sali sejmowej, otrzymują z opóźnieniem. Dlatego bardzo prosiłbym o stwierdzenie kworum, a jeżeli tak jest, o odpowiednie wydruki, żeby można było w sposób zgodny z prawem obradować. Dziękuję. Dziękuję, panie pośle. Wyprzedził pan tym wnioskiem formalnym to, co muszę zrobić oczywiście, czyli stwierdzenie kworum. Za chwileczkę odbędziemy takie głosowanie - każdy, kto jest, także zdalnie.

Czwartek był przeznaczony na cały dzień prób.

Nie wiem w jakim celu - czy po to, żeby inni w tej chwili się łączyli i żeby zablokować serwery.

Zwracam się do wszystkich państwa - także tych, którzy są w innych salach, ale również tych, którzy są poza salą plenarną - o to, żebyśmy mogli stwierdzić kworum. Jeżeli będą jakieś kłopoty, nastąpi przerwa techniczna. Bardzo proszę. Ci, co są obecni na sali, mają karty i głosują kartami. Każdy z państwa otrzymał kod, który jest kodem do zalogowania się do systemu głosowań. Oczywiście, panie pośle, będzie to trwało trochę dłużej, bo transmisja z sali posiedzeń dociera do posłów, którzy są poza salą, także z nieznacznym opóźnieniem. Biorę to wszystko pod uwagę, dlatego będziemy robić to wolniej, będziemy czekać. W tej chwili zwracam się do wszystkich państwa posłów obecnych tutaj, w innych salach i poza budynkiem sejmowym, żeby przygotować się do głosowania. Przypominam, że trzeba wcisnąć kod, który państwo otrzymaliście. To jest wasz osobisty kod do głosowań. Odczekam chwilę i za chwileczkę przystąpimy do głosowania, żeby stwierdzić kworum.

Pani poseł Katarzyna Kotala z Lewicy, tak?

Proszę państwa, klub parlamentarny Lewicy zgłasza wniosek formalny o przedłużenie posiedzenia Sejmu - na sobotę i niedzielę. Wczoraj licytowaliśmy się wszyscy w tym, że jesteśmy gotowi do pracy. Ustaw jest dużo, Polacy nie mogą już dłużej czekać na dobre rozwiązania. Proponujemy więc zostać na sobotę i niedzielę i procedować nad wszystkimi pilnie potrzebnymi ustawami, tak żeby Polacy mogli otrzymać realną pomoc. Tylko, pani poseł, to nie jest wniosek formalny, tak sformułowany, ale rozumiem pani intencję. Pani Poseł! Pani Marszałek! Ja bardzo bym prosił, żeby pani w tym szczególnym momencie obrad Sejmu dyscyplinowała takich posłów jak pan Nitras, który - kiedy nasza posłanka wygłasza wniosek formalny - przerywa i pokrzykuje. Jeżeli to się będzie działo dalej, to przerwijmy te obrady. To jest niegrzeczne. Apeluję do opozycji, całej naszej: dlaczego się kłócicie?

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Znaleźliśmy się dzisiaj w niezwykłych okolicznościach. W okolicznościach, kiedy cały świat walczy z pandemią koronawirusa. Jak bardzo nietypowe to są okoliczności, te dni i te tygodnie, niech świadczą komentarze niektórych przywódców unijnych, np. premiera Włoch, który mówi, że to jest najtrudniejszy czas od czasów II wojny światowej. Podobnie mówi kanclerz Merkel. My, Polacy, doświadczyliśmy koszmaru II wojny światowej i później w czasach komunizmu doznaliśmy również wielu cierpień, więc takich porównań nie czynimy, ale z całą pewnością to, co stało się teraz, to, co dzieje się na naszych oczach, jest największym wyzwaniem ostatnich dziesięcioleci. Dane, które napływają do nas z poszczególnych państw, instytutów, agencji ratingowych i które wskazują na perspektywy gospodarcze, są zatrważające. W Stanach Zjednoczonych właśnie podano dane dotyczące liczby osób, które zgłosiły się po zasiłek dla bezrobotnych. Otóż są to liczby największe w historii.

Dzisiaj to jest ponad 3300 tys. osób w Stanach Zjednoczonych. Te dane zatrzęsły światem i uświadomiły wszystkim, w jak trudnym położeniu dzisiaj znajduje się gospodarka globalna, w jak dramatyczny sposób wszyscy na świecie muszą dzisiaj zjednoczyć się, żeby walczyć z koronawirusem, ale też nie podejmować tego na zasadzie fałszywego wyboru, czy walczymy o zdrowie publiczne, czy walczymy, trochę w darwinistyczny sposób, o gospodarkę, bo takie głosy też dały się usłyszeć. My uważamy, że to jest błędny wybór. My uważamy, że trzeba maksymalnie spowalniać rozprzestrzenianie się koronawirusa, ale jednocześnie mamy świadomość, że dzieje się to z ogromną szkodą dla gospodarki, że dzieje się to w sposób niszczący dla gospodarki europejskiej, gospodarki polskiej. Dane, które napływają z zachodniej Europy, pokazują, że nasze działania są właściwe, często wyprzedzające. Nie mamy z tego powodu żadnej szczególnej satysfakcji, jesteśmy jedynie przekonani, że dzisiaj musimy działać szybko. Trochę tak jak przy wykryciu jakiejś groźnej bardzo choroby - jeden dzień zwłoki to ogromna różnica. Piątek czy sobota - to może być ogromna różnica. Dlatego proszę dzisiaj Wysoką Izbę, żeby wszyscy w zgodzie przyjęli ten pakiet, który przygotowaliśmy. Nasza tarcza antykryzysowa jest dobrym instrumentem na ten etap rozwoju koronawirusa i walki z wirusem w gospodarce. Musimy działać błyskawicznie, musimy działać jak najszybciej. Chcemy doprowadzić do tego, żeby te instrumenty działały już na dniach. Apeluję do przedsiębiorców, bo to w waszych przedsiębiorstwach już właściwie codziennie podejmowane są decyzje co do przyszłości. Tarcza antykryzysowa ma z jednej strony chronić miejsca pracy, z drugiej strony chronić przed bankructwami.

To potwierdzają już dzisiaj bardzo liczne instytuty, bardzo wiele badań gospodarczych i danych gospodarczych to potwierdza.

Nie trzeba być ekonomistą, żeby zdawać sobie sprawę z tego, co to może oznaczać dla gospodarki europejskiej, dla gospodarki polskiej. Prognozy dla Włoch: minus 7% to są dzisiaj już normalne prognozy, a to jest też nasz bardzo ważny partner handlowy. Dzisiaj poszarpane zostały wszystkie łańcuchy dostaw, łańcuchy produkcji.

Mamy do czynienia ze zjawiskami bezprecedensowymi.

Trzeba działać szybko. Spadki na rynkach surowców, spadki na rynkach różnych aktywów pokazują, że dzisiaj trzeba zjednoczyć się w walce ze skutkami gospodarczymi, które już toczą gospodarkę. Ten kryzys na pewno uderza w stronę popytową, podażową, konsumpcję, inwestycje, ma charakter odmienny. Wszystkie poprzednie kryzysy charakteryzowały się brakiem popytu. Ten kryzys jest inny. Musimy jednocześnie pracować nad mechanizmami ustabilizowania łańcuchów dostaw, łańcuchów produkcji, mechanizmów podaży, bo one również zostały zakłócone. To dlatego rząd Rzeczypospolitej Polskiej działa tak szybko, jak to możliwe. W 14 dni od pojawienia się pierwszego przypadku osoby chorej na koronawirusa przedstawiliśmy pierwsze założenia tarczy antykryzysowej. Nie wiem, może ktoś był na świecie odrobinę szybszy, ale jest to na pewno jedna z najszybszych odpowiedzi na to, co się dzieje wokół nas. Musimy zareagować zdecydowanie, i reagujemy zdecydowanie, tak jak dzisiaj, po kilku dniach od zaprezentowania charakterystyki naszej tarczy antykryzysowej. Potwierdzają to najsłynniejsi ekonomiści świata i instytuty badawcze, instytuty ekonomiczne. Działamy na stronę podażową, na stronę popytową. Staramy się za wszelką cenę zapobiegać bankructwom firm i zwolnieniom pracowniczym. To jest warunek sine qua non powstrzymania spirali, która później pociągnie konsumpcję i inwestycje, która może spowodować drżenie w różnych częściach gospodarki - w obszarze fiskalnym, finansowym, monetarnym, w gospodarce realnej. Dzisiaj, jak nigdy wcześniej, potrzebujemy współpracy - współpracy w ramach policy mix, mieszanki polityk, najlepszych polityk gospodarczych: polityki monetarnej, fiskalnej, regulacyjnej, w odniesieniu do gospodarki realnej. Pandemia koronawirusa, jak widzimy w kilku państwach, również u naszych przyjaciół, naszych partnerów z zachodniej Europy, powoduje istne gospodarcze, zdrowotne pandemonium. Nie chcemy doprowadzić do tego w Polsce. Bronimy się przed tym i na razie z pokorą, ale też z zadowoleniem możemy powiedzieć, że robimy wszystko co w naszej mocy, żeby tę krzywą wzrostu spowolnić. Wiele analiz pokazuje, że ta krzywa przebiega inaczej. To jest pewna iskierka nadziei. To jeszcze nie jest zwycięstwo, to jeszcze nie oznacza zwycięstwa, ale to jest, owszem, światełko w tunelu. To spowolnienie spowoduje, że nasza służba zdrowia będzie w stanie lepiej świadczyć usługi medyczne, lepiej opiekować się osobami chorymi, tak żeby nie dochodziło do sytuacji strasznych, takich sytuacji, jakie widzimy w Hiszpanii i we Włoszech, do segregacji. Chcemy za wszelką cenę tego uniknąć, chcemy przede wszystkim zdążyć na czas ze szpitalami jednoimiennymi, z nowymi miejscami w różnych szpitalach, z nowymi miejscami do kwarantanny. Dziękuję przy okazji rodakom i apeluję zdecydowanie o to, żeby wszyscy trzymali się zasad, rygorów kwarantanny i rygorów dystansowania się od siebie, żeby przestrzegali zasad sanitarnych i higienicznych. One, zdaniem epidemiologów, są krytycznie ważne po to, żeby w takiej, nazwijmy to umownie, nowej normalności wrócić do życia zawodowego w większym wymiarze, do handlu międzynarodowego. Pewnie wszyscy obserwują różne trendy. Dzisiaj trendy na rynkach, na rynkach finansowych, na rynkach oddających wartości surowców, aktywów różnego rodzaju, się załamały. Wszystkie te trendy się załamały, ale nasza odpowiedź na tym etapie jest najwłaściwsza spośród tych, jakie ktokolwiek inny wymyślił. Nasza odpowiedź, nasza tarcza antykryzysowa to ok. 10% PKB - 10% PKB składające się z różnych instrumentów. Po pierwsze i przede wszystkim, zapobieganie zwolnieniom. Drodzy pracodawcy i przedsiębiorcy, te środki, które zaoferowaliśmy.

To jest fundamentalnie potrzebne, bo ja wierzę w odbicie gospodarcze w kształcie litery V, jak mówią makroekonomiści. W najgorszym razie w kształcie litery U, ale takiej o krótkim okresie recesji, krótkim okresie spowolnienia, a to oznacza, że dobrze jest móc przechować wszystkie atrybuty, wszystkie parametry mikrogospodarcze działania waszych przedsiębiorstw w tak szerokim zakresie, jak to jest możliwe. Gospodarka to w końcu przecież również zaufanie i powiązania pomiędzy firmami, między konsumentami, obywatelami a firmami, firmami jednymi a drugimi, B2B, B2C, C2G itd., wszystkie te litery można ze sobą nawzajem mieszać. Fachowcy wiedzą doskonale, że te powiązania wymagają przynajmniej przechowania przez jakiś czas zdolności produkcyjnych i zatrudnienia w poszczególnych firmach, w poszczególnych branżach. Dla osób szczególnie dotkniętych mamy w naszej tarczy antykryzysowej rozwiązania szczególnie do tego dostosowane: pełne zwolnienie z ZUS. które wcześniej były na umowach-zleceniach, na umowach cywilnoprawnych i straciły te zlecenia. Dla wszystkich pracowników, również firm do dziewięciu osób, czyli tych najbardziej dotkniętych koronawirusem, jest zwolnienie z ZUS, jest również dodatkowy zastrzyk finansowy dla wszystkich tych firm, opisany bardzo szczegółowo w I i w II filarze. Dla osób, które są na postojowym - nie tylko dopłata 40% do wynagrodzenia, 40% średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ale również zwolnienie z ZUS.

To są pieniądze, które przekazaliśmy na politykę społeczną. Ta polityka społeczna stanowi dzisiaj bardzo ważny amortyzator. Całe 500+, również na pierwsze dziecko, utrzymujemy. To bufor społeczny dla rodzin, dla tych rodzin szczególnie dotkniętych koronawirusem, dotkniętych szczególnymi warunkami na polu gospodarczym. Oczywiście utrzymujemy również emeryturę+, także wyprawkę, również obniżkę do zera w podatku PIT dla młodych osób, tak żeby przejść przez te trudne miesiące w sposób solidarny, razem. To wszystko utrzymujemy. Jesteśmy na tym etapie przygotowani również dlatego, że doprowadziliśmy gospodarkę polską do stanu, w jakim ona wcześniej nie była, do jednego z najniższych poziomów długu publicznego.

To jest niestety przez koronawirusa rozdział zamknięty, ale to daje nam siłę, siłę budżetową, monetarną do właściwej odpowiedzi na te zmagania, które są przed nami, na ten bardzo trudny okres, który jest przed gospodarką światową, a przed gospodarką europejską dramatycznie trudny. Polska jest w lepszym położeniu, ale podchodzimy do wyzwań z ogromną pokorą. Zdaję sobie sprawę z tego, że wymaga to subtelnych, misternych powiązań pomiędzy polityką monetarną w jej różnych odsłonach, nie tylko stopy procentowe, nie tylko różnego rodzaju LTRO i działania zsynchronizowane z rynkiem, takie jakie są prowadzone, ale również, zgodnie z zaleceniami, które teraz, na dniach, są formułowane przez najlepsze instytuty badawcze, uruchomienia polityki fiskalnej. I dlatego zaproponowaliśmy jesienią zeszłego roku budżet bez deficytu. Dla nas najważniejsi są Polacy. I będziemy używać pieniędzy budżetowych do takiego stopnia, do jakiego będzie to konieczne, ale zarazem do takiego stopnia, który da nam i rynkom zewnętrznym, z którymi jesteśmy w ciągłym, codziennym dialogu, przekonanie co do stabilności naszej polityki monetarnej, polityki fiskalnej i polityki regulacyjnej. To dlatego w taki, a nie inny sposób proponujemy regulacje w odniesieniu do wymogów kapitałowych. Dlatego w taki, a nie inny sposób niezależny bank centralny zadziałał na stopie rezerwy obowiązkowej, czyli odwrotności mnożnika kreacji pieniądza. To są działania najbardziej potrzebne na ten okres. Ale zdaję sobie dzisiaj doskonale sprawę, że to w każdej godzinie zapadają decyzje w zarządach firm, tych większych, u właścicieli firm mniejszych, dotyczące reorganizacji biznesu, zwalniania pracowników bądź sprzedaży części aktywów. I chciałem zaapelować o współpracę, bo jestem przekonany, że w ciągu paru miesięcy będziemy, cała Europa, w lepszym stanie, jeśli chodzi o koronawirusa, i wtedy wygrywać będą ci, którzy będą mieli najlepiej dopasowane struktury organizacyjne, struktury biznesowe, struktury produkcji i usług do gospodarki, która przecież będzie się odradzać. Po tych wielkich spadkach w Stanach Zjednoczonych, w Unii Europejskiej, zachodniej części Unii Europejskiej handel z powrotem ruszy. Dzisiaj przedsiębiorcy wiedzą, że on jest przymrożony, mówiąc delikatnie, ale przecież handel będzie się odradzał. I dlatego tak ważne jest, by być wtedy gotowym, żeby móc wskoczyć w to miejsce. A rośnie świadomość w Unii Europejskiej. Wczoraj, tydzień temu, dwa tygodnie temu, codziennie rozmawiam z przywódcami Unii Europejskiej. Rośnie świadomość tego, że Unia Europejska musi aktywnie uczestniczyć w globalnej przebudowie struktur produkcji i powiązań produkcyjnych całego świata. I my, Polska, musimy być do tego przygotowani. Musimy być przygotowani nie tylko w tych obszarach, w których dzisiaj jesteśmy szczególnie dotknięci - wyprzedany sektor farmaceutyczny, brak wielu sprzętów - to będzie odtwarzane w całej Europie i Polska na pewno będzie w awangardzie branż, które będą odtwarzały swoje moce produkcyjne, swoje zdolności. Ale również rozmawiamy w Unii Europejskiej o tym, żeby właśnie razem, w solidarny sposób znaleźć odpowiedź na te trudne wyzwania. Niestety dzisiaj Unia Europejska nie dała jeszcze żadnego eurocenta na walkę z koronawirusem. Widać, że w takich czasach jak te, czasach bardzo trudnych, najważniejsze są państwa, państwa narodowe. No bo niestety reakcje Unii Europejskiej są, może powiem: są, jakie są, każdy może je zaobserwować, bo o tym, że to nie są nowe pieniądze. A więc to pozostaje poza jakąkolwiek wątpliwością. Jednak wierzę, że w sposób spóźniony, po odpowiedniej stymulacji. Ona była również wczoraj, mówili o tym premier Hiszpanii i premier Włoch, premierzy Grupy Wyszehradzkiej, wraz ze mną, i kilku innych krajów, bardzo mocno podnosząc, że jeżeli Unia Europejska ma utrzymać zaufanie obywateli, musi odpowiedzieć na to w sposób adekwatny.

Jaka jest odpowiedź Unii Europejskiej jako całości? Poczekamy. Mam nadzieję, że będzie. Na razie odpowiedź jest po stronie państw narodowych. Warto, żeby wszyscy to wiedzieli, warto też, żeby każdy to sobie uświadomił - że walka z tymi przeciwnościami losu zarówno od strony mechanizmów podażowych, popytowych, jak i fiskalnych odbywa się poprzez budżety poszczególnych państw członkowskich. Oprócz działań osłonowych na rynku pracy, o których powiedziałem, oprócz wielu działań, które są w naszym tzw. II filarze, gdzie uruchamiamy pieniądze gwarancyjne i pieniądze bezpośrednie - i to są również realne pieniądze, dziesiątki miliardów złotych, co najmniej 70 mld zł na utrzymanie płynności w firmach, na bezzwrotne pożyczki, na zwrotne pożyczki, na leasing operacyjny, na kredyty, na płynność, kredyty obrotowe, kredyty bieżące, kredyty w rachunku bieżącym, ale również na bezpośrednie dopłaty po to, żeby przedsiębiorcy z branż takich jak turystyczna, gastronomiczna, transportowa, logistyczna, handlowa - wielka, bardzo ważna branża - nie pozostali sami i oni nie pozostaną sami. My proponujemy w ramach tarczy antykryzysowej szereg rozwiązań dostosowanych również do poszczególnych branż. Dziękuję za wszystkie refleksje, za możliwość usprawnienia tego pakietu na tym etapie, na jakim on dzisiaj został zatwierdzony. To nie jest ostatnie słowo, ba, jestem przekonany, że to jest dopiero pierwsza nasza odpowiedź. Będziemy dostosowywać się do potrzeb rynku, będziemy obserwować. Codziennie spotykamy się na forum gospodarczym, na forum głównych aktorów sceny gospodarczej.

Chcę wszystkich państwa i wszystkich rodaków zapewnić, że nie zostawimy was samych. Państwo polskie idzie tą wąską granią, gdzie po jednej stronie mamy bezrobocie, bankructwa firm - i chcemy im zapobiegać, używając najmocniejszych mechanizmów fiskalnych i monetarnych, jakie są dostępne - ale po drugiej stronie mamy wiarygodność naszych instrumentów wobec świata zewnętrznego. Wczoraj słyszałem, tutaj siedząc, pewien koncert życzeń. Drodzy państwo, drodzy przedstawiciele opozycji, wiecie, że jestem otwarty na dialog. W ostatnich kilku tygodniach osobiście spotykałem się z wami wielokrotnie, kilkukrotnie w formacie bezpośrednim, i dodatkowo kilka razy w formacie Rady Bezpieczeństwa Narodowego zwoływanej przez pana prezydenta. Wiecie doskonale, że potrafimy słuchać, wykorzystywać pewne pomysły, które są dobre, ale jednocześnie zdajcie sobie sprawę z tego, że dzisiaj wiarygodność na rynkach, na rynkach globalnych, finansowych, decyduje o zdolności do przeprowadzania jakichkolwiek działań gospodarczych. Są państwa, które już zbankrutowały, których dług nie został wykupiony. To państwa wysoce zadłużone. Nasz wzrost gospodarczy był zrównoważony, dług publiczny spadał do PKB, dług prywatny i dług przedsiębiorstw był niższy od średniej. W związku z tym mamy pewne bufory do uruchomienia i uruchamiamy je. To bardzo ważne filary w naszej tarczy antykryzysowej, które mają na celu zrestartowanie gospodarki i inwestycji, natychmiast jak odbudowane zostanie zaufanie w podstawowej, elementarnej warstwie - czyli mam nadzieję, że już za kilka tygodni, że już wkrótce. Najpierw trzeba zdusić, opanować koronawirusa. Chiny nie są państwem demokratycznym. Udało się to w Korei, udało się to w Japonii, udaje się to na Tajwanie. Tamte państwa również mają inną kulturę polityczną, inną kulturę relacji społecznych, ale my chcemy wykorzystywać i wykorzystujemy tamte doświadczenia. To jest nasza metoda walki z tą globalną pandemią, która jest pierwszym takim wyzwaniem zdrowotnym dla świata - pomijając oczywiście wojny - od 1918 r., od grypy hiszpanki. COVID-19 to wielki kryzys zdrowotny, który w wielu krajach świata już przekształcił się w głęboki kryzys gospodarczy. My nie jesteśmy samotną wyspą, jesteśmy współzależni od reszty świata. Mamy bardzo otwartą gospodarkę.

Dzisiaj, kiedy te branże stają, kiedy Volkswagen, Opel, Fiat, Mercedes, BMW wstrzymują produkcję, polscy dostawcy części również wstrzymują produkcję. My na ten czas, na te kilka tygodni, może na miesiąc, dwa, trzy - mam nadzieję, że nie dłużej, i wierzę w to, że nie dłużej, jak patrzę na sygnały płynące z różnych stron świata - przygotowaliśmy najwłaściwsze rozwiązanie gospodarcze i to jest nasza tarcza antykryzysowa. Dzisiaj również obywatele chcą od nas zapewnienia spokoju i pewności co do ich oszczędności. Stąd filar zapewnienia tego bezpieczeństwa, który zapewniają KNF, Ministerstwo Finansów i przede wszystkim również Narodowy Bank Polski. Nie dajemy sektorowi bankowemu w sensie dotacji ani złotówki. Podkreślam to, ponieważ pojawiły się liczne fake newsy. Rozumiem walkę polityczną, ale dzisiaj mówienie prawdy jest ważniejsze, bo jeden fake news może spowodować bardzo duże szkody w całej gospodarce. Apeluję zatem o to, żeby działać razem, działać wspólnie. To jest sprawa arcypoważna. Mamy przekonanie, że na tym etapie nasza odpowiedź jest najbardziej adekwatna.

Ważne jest, aby zrobić to niemal natychmiast, bo każdy dzień zwłoki oznacza dziesiątki tysięcy bezrobotnych.

Dlatego bardzo proszę Wysoką Izbę, mając na uwadze powagę sytuacji, w jakiej się znajdujemy, żeby nie toczyć jałowych sporów, nie tworzyć u rodaków wrażenia, że można rozkręcić koncert życzeń, że każde 10, 50 mld zł każdy może położyć na stole. Proszę wejść z nami w dialog, dialog, w którym to wam pokażemy, jeżeli ktoś nie ma dostępu, bo przecież właściwie wszystkie dane fiskalne, monetarne są dostępne, można je poprzeliczać i wszystko widać.

Dlatego bardzo proszę Wysoką Izbę, głosujmy szybko, głosujmy zgodnie nad tą arcypoważną sprawą w sytuacji, w jakiej jesteśmy, bo od tego zależy przyszłość polskiej gospodarki i przyszłość Polaków. Dziękuję, panie premierze. Proszę o zabranie głosu ministra rozwoju panią Jadwigę Emilewicz i przedstawienie uzasadnienia projektów ustaw zawartych w drukach nr 299, 299-A i 302. Bardzo proszę, pani minister. Panie i Panowie Posłowie! Tak jak powiedział pan premier, mam przyjemność przedstawić państwu ustawę o zapobieganiu rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, i tak jak powiedział pan premier, nad tą ustawą pracowali wszyscy ministrowie w naszym rządzie. Konsultowaliśmy się ze stroną pracowników i pracodawców, rozmawialiśmy codziennie z wieloma przedstawicielami wielu branż. Zdajemy sobie doskonale sprawę, w jakiej sytuacji znajduje się dzisiaj polska gospodarka. Jestem przekonana, podobnie jak pan premier, że dla pokolenia takiego jak moje, pokolenia wychowanego w wolnej Polsce pandemia i jej społeczne konsekwencje będą doświadczeniem pokoleniowym. Dla części z państwa posłów takim doświadczeniem były na pewno „Solidarność”, stan wojenny i budowanie wolnej Polski na początku lat 90. Dla nas z całą pewnością te wydarzenia, które są dzisiaj, i ich konsekwencje będą takim doświadczeniem. Mam nadzieję, że zdamy egzamin z tego doświadczenia w podobny sposób, jak zrobili to nieco starsi państwo posłowie.

Niech mi chociaż będzie wolno zauważyć, że największe koszty zapewne poniesie pokolenie tych osób, które nie mają jeszcze ustabilizowanej sytuacji zawodowej i materialnej, dzisiejsi 20-, 30-, a może także 40-latkowie. Rozwiązaniami, które proponujemy, staraliśmy się objąć wszystkich pracowników i pracodawców, ale oczywiście same ustawy nie wystarczą. Będziemy znowu, jak 40 lat temu, próbować budować solidarność. Będziemy tej solidarności bardzo potrzebować, solidarności młodszych ze starszymi, solidarności miedzy pracodawcą a pracownikiem, solidarności pomiędzy przedstawicielami administracji a wszystkimi obywatelami. W zakresie zdrowia wyrazem solidarności jest dzisiaj dystans, ten dystans jednak paraliżuje naszą gospodarkę. Dlatego przygotowaliśmy rozwiązania, które mają sprawić, że przez ten trudny okres przeprowadzimy zarówno pracowników, jak i pracodawców w miarę możliwości, jak tylko to będzie możliwe, suchą stopą. Tak jak już wspomniał pan premier, tworzymy elastyczne ramy służące temu, aby tę pomoc dostarczać.

Dlatego jednym z elementów wprowadzanych w przedłożonej ustawie jest stworzenie Funduszu COVID-19. To jest nowy fundusz, którego dysponentem będzie prezes Rady Ministrów. Środki tego funduszu będą mogły być dystrybuowane do innych funduszy, do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Funduszu Pracy, tam gdzie w danym momencie będą potrzebne, ponieważ nie zabraknie środków na udzielanie pomocy tym wszystkim, którzy spełniają dzisiaj kryteria, aby tą pomocą mogli zostać objęci.

One też będą mogły teraz skorzystać z takich świadczeń. Zmieniamy również zakres tej pomocy dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Wprowadzamy rozwiązania z zakresu ochrony miejsc pracy, jak mówił pan premier. Tutaj proponujemy szeroki wachlarz ułatwień. Dla firm, zarówno małych, jak i większych, znosimy reżim pomocy de minimis, pomocy publicznej, znany z czasów przedwirusowych, a zatem nie mamy żadnego limitu pomocy publicznej w tym zakresie. Oferujemy dwa rodzaje rozwiązania.

W ramach tego postoju może zredukować czas pracy wszystkich pracowników do wymiaru połowy etatu, tej połowy, która jednak nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie.

Jeśli przedsiębiorstwo spowalnia, ale może świadczyć usługi, może prowadzić, kontynuować, choć w zredukowanym wymiarze, działalność produkcyjną, wówczas przedsiębiorca może redukować czas pracy swoich pracowników o 20%, do wymiaru 0,8 etatu. I wówczas także fundusz świadczeń gwarantowanych pokryje połowę wynagrodzenia, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, czyli do kwoty ok. 5 tys. zł. Połowę tej części pokryje fundusz świadczeń gwarantowanych - i tutaj znowu wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Drugą część będzie pokrywał pracodawca. To bardzo konkretne i bardzo silne wsparcie, które w przypadku postojowego obniża koszty działania, działalności firmy o ok. 80%. Te rozwiązania, tak jak powiedziałam, są powszechne. Mogą z nich korzystać zarówno małe firmy - do 10, 20, 30, 50 pracowników - jak i wszystkie firmy duże, które nie mieszczą się w kryterium małego i średniego przedsiębiorcy. Te duże firmy, które korzystały z pomocy publicznej czy to w zwolnieniach podatkowych, czy w bezpośrednich grantach, czy korzystając z mechanizmów specjalnych stref ekonomicznych - ta pomoc udzielana w poprzednich latach się nie sumuje - dziś mogą korzystać z tej pomocy dla podtrzymania pracowników i podtrzymania stanu. Ułatwiamy i uelastyczniamy możliwość korzystania z tych instrumentów, tzn. przedsiębiorca może łącznie korzystać i z jednego, i z drugiego, może część pracowników wysłać na postojowe, a części obniżyć wynagrodzenie, pozostawiając ich w pracy. Taki pracodawca może także skorzystać z prolongaty zarówno składek na ubezpieczenia społeczne, jak i wszystkich swoich obowiązków podatniczych. Dotychczas mógł to robić, ale musiał ponieść z tego tytułu opłatę prolongacyjną. My tę opłatę znosimy. O odroczenie bądź układ ratalny będzie można zwrócić się na bardzo prostym, 1-stronicowym formularzu. One wszystkie będą dostępne już w przyszłym tygodniu i dla pracowników, i dla pracodawców. Podobnie właściwe naliczenia na podatki - również będzie mogło to odbyć się na podstawie bardzo prostego oświadczenia, które także będzie dostępne już w przyszłym tygodniu. Jednocześnie w tym okresie oferujemy mikrofirmom, tak jak wspomniał pan premier, zniesienie składek na ubezpieczenia społeczne. Firmy zatrudniające od jednego do dziewięciu pracowników będą mogły skorzystać ze zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne, jeśli ich obroty spadły o ok. 50% w miesiącu poprzedzającym. Właściciel takiej firmy, który jest bardzo często samozatrudniony, również nie będzie musiał płacić składek na ubezpieczenia społeczne, jeśli jego przychody nie przekroczyły trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia, czyli dziś jest to 15 600 zł. Na jeden kwartał znosimy także obowiązki składek na ubezpieczenia społeczne dla tych ubezpieczonych w rolniczym systemie ubezpieczeń społecznych.

One także będą dostępne w dniu wejścia w życie tej ustawy. Dla pracodawców, którzy będą korzystać czy to z rozwiązania postojowego, czy też z rozwiązania dotyczącego obniżonego wymiaru pracy, uelastyczniamy także możliwości rozliczania czasu pracy. Będą mogli wykorzystywać to w okresie już popostojowym, wówczas kiedy wrócą do pełnego wymiaru pracy, w większym stopniu korzystać z pracowników, i skróci się czas odpoczynku dla pracowników. Jest to - co chciałabym podkreślić - rozwiązanie, które wypracowaliśmy ze stroną społeczną. Strona społeczna, przedstawiciele wszystkich związków zawodowych, rozumiejąc powagę sytuacji, zgodzili się na te rozwiązania, na które przez wiele lat nie wyrażali zgody. Rozumieją, że ta elastyczność jest dzisiaj warunkiem utrzymania miejsc pracy. Ta ustawa wprowadza także szereg ułatwień biurokratycznych. Wiążą się one chociażby z wydłużeniem wielu terminów administracyjnych. Jeżeli komuś kończy się termin ważności takich badań, będzie on w czasie trwania epidemii wydłużony w sposób automatyczny. Wydłużamy także okres ważności zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych.

Mamy także w tym pakiecie specyficzne branżowe rozwiązania dotyczące sektora szeroko związanego z sektorem kultury. Dla tych, którzy dzisiaj nie mogą z powodu zakazów i ograniczeń w ruchu prowadzić swojej działalności, w dyspozycji ministra kultury i dziedzictwa narodowego pozostaje fundusz, którym minister będzie mógł dysponować w sposób swobodny po to, aby podtrzymać tę aktywność w czasie, kiedy ona w trybie normalnym nie może być prowadzona. To ta branża, która w pierwszej kolejności ucierpiała z powodu rozprzestrzeniania się wirusa. Wprowadzamy zatem rozwiązanie. Jak państwo wiedzą, dziś, kiedy impreza turystyczna, z której chcieliśmy skorzystać, jest anulowana przez organizatora, możemy ubiegać się o zwrot kosztów w terminie do 14 dni od dnia anulowania wydarzenia. My wydłużamy ten termin do 180 dni - to są takie rozwiązania, jakie zostały przyjęte również w ostatnich tygodniach w kilku państwach członkowskich - oraz dajemy możliwość zwrotu kosztów tego wydarzenia nie tylko w formie gotówkowej, ale także w formie vouchera na poczet nowego, innego wydarzenia.

Wprowadzamy także rozluźnienia w zakresie wymogów wynikających z Prawa zamówień publicznych. Wiele inwestycji, realizacji nie będzie mogło być dokończonych w terminach wynikających z umów właśnie ze względu na trwający stan epidemii.

Przedłużamy także i adresujemy rozwiązania związane z rynkiem pracy. W sposób automatyczny przedłużeniu ulegają wizy i pozwolenia na pobyt, pozwolenia na pracę w czasie trwania stanu epidemii oraz w okresie 60 dni po jego zakończeniu. To jest bardzo ważny element, na który zwracali nam uwagę pracodawcy. Jednocześnie wprowadzamy rozwiązania adresowane do tych, którzy wynajmują powierzchnie w sklepach wielkopowierzchniowych, galeriach, które dzisiaj są zamknięte, w obiektach handlowych. Wprowadzamy rozwiązanie, zgodnie z którym. Na mocy dzisiejszego prawa wiemy, że stan, w którym dzisiaj jesteśmy, zwalnia z obowiązków prawnych najemców. Tymi obowiązkami jest płatność czynszu. Wprowadzamy dodatkowo takie elementy, które sprawią, że po zakończeniu tego stanu w sposób automatyczny będą wygasać podpisane dzisiaj umowy i najmujący będą podpisywać nowe umowy. Na mocy tych nowych umów wydłużamy pas startowy i te pierwsze miesiące będą obłożone niższym czynszem niż przed czasem wirusa. Dajemy w ten sposób szanse na przetrwanie tym branżom i tym firmom, które dzisiaj nie mogą prowadzić swojej działalności. W zakresie nowych obowiązków, które miały wejść w życie w tym roku, znosimy je bądź przesuwamy część z nich. Przesuwamy wejście w życie bazy danych o odpadach, nowych obowiązków administracyjnych dla wszystkich przedsiębiorców. Przesuwamy ten termin na koniec roku. Wprowadzamy także elastyczne formy zmiany planów finansowych w instytucjach niezbędnych, które mierzą się dzisiaj z problemami związanymi z rozprzestrzenianiem się wirusa. Są to takie instytucje jak Agencja Rezerw Materiałowych czy KOWR, które będą mogły w sposób swobodny zmieniać plany finansowe bez konieczności notyfikowania ich przez Komisję Finansów Publicznych. Tylko w ten sposób będziemy mogli aktywnie odpowiadać na potrzeby dzisiejszych czasów. W zaprezentowanych przez nas rozwiązaniach są także szczególne rozwiązania dotyczące pomocy de minimis, pomocy znanej większości firm w Polsce. Jest to pomoc pożyczkowa, której gwarantem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Dotychczas ten instrument był ograniczony do 60%, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego gwarantował pożyczkę do wysokości 60% jej wielkości. My podnosimy tę gwarancję do 80% i zwiększamy wolumen, z którego może firma skorzystać, z 200 do 800 tys. euro. Dystrybutorem tych pożyczek są banki komercyjne. Są to, możemy powiedzieć, tanie i proste pożyczki obrotowe, które pozwolą firmom przetrwać ten trudny czas. Całość tak naprawdę ryzyka zostaje tutaj przeniesiona na Bank Gospodarstwa Krajowego. Przedsiębiorca nie musi zatem dostarczać i spełniać bardzo wysokich wymogów wynikających z Prawa bankowego. Do całości rozwiązań, które proponujemy, dołączamy także... do filarów, o których wspomniał pan premier, tych filarów inwestycyjnych. Tego filaru dotyczy ustawa zmieniająca ustawę o systemie instytucji rozwoju. W ramach systemu instytucji rozwoju uruchamiamy dwa instrumenty. Jeden z nich to: w Agencji Rozwoju Przemysłu zostanie uruchomiony instrument wsparcia branży transportowej. Polska jest tym państwem, które stanowi najwięcej usług transportowych w całej Europie.

Większość. Mamy 278 tys. ciężarówek, których właścicielami są zarówno duże firmy, jak i gros z nich, 25% tych firm to są firmy mikro i małe. Większość tych ciężarówek to są ciężarówki leasingowane. Dzisiaj spłata rat leasingowych jest ogromnym wyzwaniem dla tych firm, dlatego w Agencji Rezerw Materiałowych utworzony zostaje specjalny fundusz w wysokości 1700 mln zł, z którego to funduszu będą finansowane przez 15 miesięcy raty leasingowe dla firm, które dzisiaj cierpią z powodu koronawirusa. W ustawie, zmienionej ustawie o systemie instytucji rozwoju zostaje wprowadzona także możliwość utworzenia nowego funduszu. Fundusz, który będzie dokapitalizowany kwotą 7 mld zł i w przypadku którego polski fundusz rozwoju będzie mógł w sposób elastyczny wchodzić udziałowo, podnosić kapitały na warunkach innych niż te tradycyjne, znane z Prawa bankowego, gdzie ocena ryzyka podmiotu będzie oczywiście znacznie inna, będzie uwzględniała sytuację, w jakiej znajdują się firmy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Niecierpliwią się państwo w tym tygodniu z tego powodu, że dostarczaliśmy ją państwu do dyskusji późno. Pomimo że pracowaliśmy nad nią nieustannie przez wiele, wiele godzin w ostatnich dobach, spotykaliśmy się z państwem, pokazując wersje robocze. Jesteśmy otwarci, bo zależy nam bardzo na tym, aby ta ustawa była, tak jak powiedziałam, projektem solidarnościowym, także projektem, który połączy nas, koalicję i opozycję, ponieważ nie robimy tego jako cel polityczny, robimy tę ustawę, przygotowujemy te rozwiązania, ponieważ one mają być dobre dla Polski. Nigdy tak. W całej historii Polski zawsze mamy takie doświadczenie, że mobilizujemy się zawsze w czasach kryzysu. Ja mam nadzieję, że z tego kryzysu będziemy, w czasie tego kryzysu będziemy nie tylko zmobilizowani ponad podziałami, ale także wyjdziemy z niego wzmocnieni. Szanowni Państwo! Dziękuję, pani minister. Teraz proszę podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia pana Janusza Cieszyńskiego o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy zawartego w drukach nr 301 i 301-A. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ja bym chciał zacząć od podziękowań, dlatego że nad tym projektem pracowaliśmy wspólnie, pracowaliśmy, wymienialiśmy się uwagami z przedstawicielami wszystkich klubów parlamentarnych, tak że moje podziękowania kieruję do pana posła Kuleszy, do pana przewodniczącego Kosiniaka-Kamysza, do pana marszałka Tyszki, do pana Darka Standerskiego z Lewicy, do pana ministra Suskiego, do wszystkich państwa, którzy w tych konsultacjach wzięli udział, i oczywiście do pana ministra Schreibera, który pomógł nam to skoordynować wraz z panią minister Emilewicz. System ochrony zdrowia wymaga pewnych dostosowań, wymaga dostosowań, które wynikają, po pierwsze, z tego, że mamy zupełnie ekstraordynaryjną sytuację, a po drugie, ze względu na to, że mamy taką konstrukcję przepisów, która pewne rzeczy na nas wymusza, pewnych rzeczy nie pozwala nam robić w sposób elastyczny. I jeśli chodzi o to, co zalecamy wszystkim obywatelom wtedy, kiedy mówimy o zwalczaniu koronawirusa, czyli ten zdrowy rozsądek, czasami te przepisy, które obecnie obowiązują, nam tego zdrowego rozsądku bez drobnych zmian nie pozwalają zastosować. Po pierwsze, chciałem tak podsumować, zmieniamy 14 ustaw, ustaw, które regulują praktycznie każdy element funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. I to jest kolejna tura zmian po tych najpilniejszych, które już zostały wprowadzone w ramach tej specustawy, która została przyjęta przez Sejm kilka tygodni temu. I chciałbym powiedzieć krótko o tych zmianach. Po pierwsze, zawieszamy egzaminy dla osób wykonujących zawody medyczne. Jeżeli ktoś zdał egzamin pisemny i czeka na ten egzamin ustny, to jeżeli nie będziemy w stanie go w określonym czasie przeprowadzić, to taka osoba, taki lekarz będzie miał ten egzamin zaliczony, czyli dopuścimy do wykonywania tych zawodów, wobec których nie jesteśmy w stanie tej drugiej ustnej części egzaminu przeprowadzić. Ograniczamy też, zawieszamy obowiązki sprawozdawcze wobec Narodowego Funduszu Zdrowia, te, które racjonalnie możemy teraz ograniczyć, ponieważ to jesz czas, szanowni państwo, na to, żeby nawet kosztem pewnych rzeczy, z których korzystają pacjenci, takich jak np. informacje o najbliższym wolnym terminie, po prostu na ten czas z tego zrezygnować. Wrócimy do tego, wrócimy do tych funkcji, z których na co dzień pacjenci korzystają, wtedy kiedy sytuacja się unormuje. Ustawy narzucają także obowiązkowe kontrole w laboratoriach diagnostycznych, stacjach krwiodawstwa i innych instytucjach ochrony zdrowia. My te kontrole także na ten moment zawieszamy i zawieszamy także funkcjonowanie instrumentu oceny inwestycji w ochronie zdrowia dla tych inwestycji, które są realizowane w związku ze zwalczaniem koronawirusa. Wiemy, że prawie 100 mln zł z rezerw ministra spraw wewnętrznych trafiło do wojewodów na niezbędne zakupy. Oczywiście ocena celowości jest bardzo istotna, ale teraz jest czas na to, aby wszystkie takie potrzeby realizować jak najszybciej.

Przede wszystkim przewidujemy możliwość włączenia do systemu lekarzy stażystów, pielęgniarek, które wracają po 5 latach lub więcej niewykonywania zawodu, osób z kursem pierwszej pomocy, które będą mogły wesprzeć pracę systemu ratownictwa medycznego.

To nie jest tak, że wprowadzamy jakieś zmiany, jak to się kolokwialnie mówi, na żywioł, tylko wprowadzamy je w taki sposób, żeby z tych zasobów, które możemy szybko pozyskać, móc skorzystać, ale bez jakiegokolwiek pogorszenia opieki nad pacjentami. Oprócz tego poszerzamy katalog podmiotów, którym minister zdrowia na podstawie specustawy będzie mógł wydawać polecenia. Rozszerzamy go o podmioty samorządowe i rozszerzamy to o możliwość wprowadzenia na czas stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego pełnomocnika ministra, który na ten okres przejmie zarządzanie szpitalem. Tego pełnomocnika powołuje minister spośród osób, które muszą spełniać takie same wymogi jak obecnie kierujący podmiotami leczniczymi.

Po zakończeniu tego okresu, po ustaniu stanu epidemii wraca osoba, która do tej pory zarządzała.

To jest niezwykle istotne, ponieważ wiemy, że zakażenia poziome mogą stanowić bardzo duże zagrożenie dla systemu ochrony zdrowia. To są sytuacje, które wystąpiły w innych krajach, i to są sytuacje, których w Polsce musimy uniknąć, tak aby system ochrony zdrowia przez cały ten czas funkcjonował sprawnie i żeby później, kiedy ta sytuacja się unormuje, wrócił do pilnej obsługi pacjentów, także tych, którym obecnie, ze względu na ryzyko zarażenia koronawirusem, odwołujemy planowe zabiegi. Oprócz tego ograniczamy katalog osób zwolnionych ze skierowania do pracy przez wojewodę.

Ta poprawka sprawia, że takie skierowanie nie będzie mogło dotyczyć kobiet w ciąży, osób wychowujących dzieci do lat 14, wychowujących dzieci niepełnosprawne lub dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jeśli chodzi o pary, które wychowują starsze dzieci, skierowanie będzie mógł otrzymać tylko jeden rodzic.

Wprowadzamy możliwość dyżurowania dla innych zawodów pracujących w ochronie zdrowia. Wprowadzamy też lepsze mechanizmy egzekucji obowiązków, egzekwowania cen maksymalnych leków i innych produktów medycznych. Przypomnę, że to są mechanizmy, tak samo jak mechanizm reglamentacji produktów leczniczych wydawanych w aptekach, których do tej pory nie zastosowaliśmy. To są mechanizmy, które wprowadziła poprzednia specustawa. To są mechanizmy, które pozwolą nam - dzięki temu, że monitorujemy cały czas stany magazynowe, że monitorujemy, ile jest wydawanych leków, jeżeli widzielibyśmy zagrożenie dla bezpieczeństwa lekowego polskich pacjentów - wprowadzić pewne ograniczenia, których na szczęście na ten moment wprowadzać nie musieliśmy. Oprócz tego wprowadzamy ułatwienia dla farmaceutów. Zgodnie z postulatami Polskiego Stronnictwa Ludowego, zgodnie z tym, co ustaliliśmy podczas naszego spotkania, wprowadzamy możliwość wystawiania przez farmaceutów refundowanych recept farmaceutycznych dla siebie i swojej rodziny oraz wydawania recept farmaceutycznych także wtedy, kiedy nie ma nagłego pogorszenia stanu zdrowia, tak jak to było do tej pory. To jest postulat, który od wielu, wielu lat wysuwało środowisko farmaceutyczne, a teraz, kiedy rola aptek jest jeszcze większa niż zwykle - przypomnę, że w tym rekordowym tygodniu polskie apteki odwiedziło 21 mln pacjentów, czyli kilkadziesiąt procent więcej niż standardowo - chcemy, żeby farmaceuci mieli dodatkowe uprawnienia i żeby w tej trudnej sytuacji mogli jeszcze lepiej pomóc swoim pacjentom. Upraszczamy także zasady udostępniania i tworzenia rezerw strategicznych na potrzeby ministra zdrowia. To jest mechanizm, który na pewno pozwoli jeszcze lepiej i szybciej dostarczyć środki ochrony indywidualnej do placówek ochrony zdrowia. Upraszczamy też dostarczanie decyzji o kwarantannie i hospitalizacji oraz o nowej instytucji, którą jest wprowadzenie izolacji w warunkach domowych.

Jeżeli nie ma konieczności hospitalizacji, to nie ma potrzeby, aby taki pacjent zajmował łóżko w szpitalu, może on spokojnie dochodzić do zdrowia w domu. Wprowadzamy także uproszczenie, jeżeli chodzi o prowadzenie dokumentacji, i wprowadzamy narzędzia cyfrowe. Szanowni państwo, to jest taki moment, kiedy widzimy, że inwestycja, strategia, którą przyjęliśmy w zakresie informatyzacji ochrony zdrowia: e-recepty, e-zwolnienia, przygotowania do wprowadzenia e-skierowań, e-dokumentacji, dzisiaj się zwraca. Myślę, że wszyscy to widzą. Jeżeli chodzi o teleporady, rodzinni lekarze podstawowej opieki zdrowotnej piszą do nas, że dzisiaj na kilkadziesiąt wizyt w ciągu dnia dwie, trzy są realizowane stacjonarnie.

Wprowadzamy taką możliwość, aby każdy, kto chciałby np. dlatego, że jest poddany kwarantannie jako lekarz czy jako pielęgniarka, udzielać takich teleporad, będzie mógł to robić. Udostępnimy taką platformę, która będzie umożliwiała wideokonsultacje, a w ramach tego wystawienie recepty, zwolnienia i wspieranie swoich pacjentów wtedy, kiedy ze względu na to, że zostaliśmy poddani kwarantannie, nie będziemy mogli im udzielać świadczeń w normalny sposób. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadza specjalną aplikację, która będzie nas wspierała przy monitorowaniu osób objętych kwarantanną.

Takim narzędziem jest ta aplikacja i ta ustawa daje nam możliwość wprowadzenia jej jako obligatoryjnego narzędzia. Oszczędzimy czas pracy funkcjonariuszy, którzy już dzisiaj wykazują wielkie zaangażowanie we wsparcie systemu ochrony zdrowia w walce z koronawirusem. Sejm ustalił, że w łącznej dyskusji nad tymi punktami porządku dziennego wysłucha 15-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Proszę.

Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec omawianych projektów, które nazwaliśmy gospodarczą tarczą antykryzysową.

Pandemia koronawirusa zmieniła nasze życie, zmieniła też nieco nasze społeczeństwo. Można powiedzieć, że rzeczywiście historia pisze się na naszych oczach, ale kiedy uświadomimy sobie, kiedy mamy w pamięci, że pokolenie naszych pradziadków walczyło pod zaborami o wolną Polskę, że pokolenie naszych dziadków walczyło w straszliwej wojnie i musiało przeżyć komunizm, że nasi ojcowie walczyli o wolną Polskę, zrzucając jarzmo komunizmu, to możemy być przekonani, i jestem przekonany, o tym, że także z tej trudnej walki, która nas czeka, wyjdziemy zwycięsko. Wysoka Izbo!

W takich sytuacjach sprawdzian stoi przed rządzącymi. Patrzę na pana ministra Mariusza Błaszczaka. Myślę, że udało się to zrobić, udało się pokazać, że państwo ma sprawstwo i że państwo nie zawodzi swoich obywateli. Gospodarcza tarcza antykryzysowa jest także taką odpowiedzią, bo owszem, możemy powiedzieć dziś, że podejmowaliśmy szybko bardzo ważne decyzje, że ograniczyliśmy imprezy masowe już po 6 dniach od pojawienia się pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce, że zamknęliśmy szkoły po 8 dniach, zamknęliśmy granice po 11 dniach, kilkakrotnie szybciej niż wszystkie inne państwa w Europie. Podejmowaliśmy, rząd podejmował decyzje dobre i trafne. Ale, szanowni państwo, są tacy ludzie, są tacy politycy w Europie, którzy mówili, przedstawiali dane, że tyle musi zachorować, a tyle niestety musi umrzeć i tak musi być. Nie, takie podejście jest nam absolutnie obce. Takie podejście dla rządu i dla Prawa i Sprawiedliwości jest nie do zaakceptowania. Trzeba walczyć o każde ludzkie życie i z tej drogi nigdy nie zejdziemy.

Wódz naczelny na niego spojrzał i zapytał, czy na ochotnika chce być jednym z tych 10.

Ale oprócz walki o zdrowie, oprócz walki o życie Polaków, którą toczą dzisiaj we wspaniały sposób także polscy lekarze, cała ochrona zdrowia, pielęgniarki, ratownicy medyczni, tej walki, za którą musimy im podziękować, stoimy także przed wielkim wyzwaniem, przed wielkim wyzwaniem kryzysu gospodarczego. Odpowiedzią na to są projekty ustaw, które dzisiaj przedstawiamy Wysokiej Izbie i o których dzisiaj rozmawiamy w Wysokiej Izbie. Szanowni Państwo! To jest, można powiedzieć, rzeczywiście taki rak, który toczy gospodarkę, i to gospodarkę całego świata. Polacy dziś mają prawo oczekiwać, że rząd nie pozostanie bierny. Mają prawo oczekiwać, że nie usłyszą ze strony przedstawicieli swojego rządu takich słów pogardliwych, jak nieraz słyszeli, że rząd się sam wyżywi - tak mówił jeden z komunistycznych aparatczyków w latach 80.

Polacy mają prawo dziś oczekiwać od rządu realnych działań.

Wysoka Izbo!

Tarcza służy nam do obrony. Dzisiaj chciałbym także zaapelować do parlamentu, zaapelować o tę jedność i o to, byśmy, wspólnie działając, mogli przyjąć tę ustawę, zaapelować do samorządowców o to, aby byli także w stanie pomóc swoim przedsiębiorcom lokalnym, zaapelować wreszcie do przedsiębiorców, byśmy wspólnie z nimi mogli ochronić miejsca pracy dla Polaków. Wysoka Izbo! Często słyszymy różne propozycje, bo ten cały katalog jest naprawdę bardzo obszerny i przemyślany, ale często też pada pytanie: No dobrze, ale co dla mnie, gdy jestem w takiej sytuacji, a co dla mnie, gdy jestem w innej sytuacji? Proszę zwrócić uwagę, że dla każdego przedsiębiorcy i dla każdej grupy są jakieś rozwiązania. Nie zapomnieliśmy o osobach, które są na umowach cywilnoprawnych. Dla nich przynajmniej to podstawowe świadczenie zostało tutaj zawarte. Nie zapomnieliśmy o osobach, które są samozatrudnione, które są na karcie podatkowej, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, które często stanęły w sytuacji dramatycznej.

Mamy propozycje dla mikroprzedsiębiorców. Dla nich również jest to rozwiązanie z ZUS-em. Po to, żeby właśnie ratowali miejsca pracy, żeby zdecydowali się ich utrzymać na rynku. Mamy wreszcie obniżenie o 90% czynszów najmów w lokalach w galeriach handlowych, które zostały naszą decyzją zamknięte. Mamy rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku. To są niezwykle ważne, konkretne propozycje. Te propozycje są też dla całego sektora małych i średnich przedsiębiorstw. To ten 40-procentowy dodatek do pensji, to otwarte linie kredytowe, to wakacje podatkowe, to refinansowanie umów leasingowych, tak jak mówiła pani minister, dla całej branży transportowej, przecież Polska jest tutaj potęgą - 27% całego rynku Unii Europejskiej to nasze firmy transportowe, nasi przedsiębiorcy. To wsparcie dla branży turystycznej, choćby przedłużenie terminu na zwrot wpłat klienta z 14 na 180 dni, to gwarancje de minimis z BGK, to dopłaty do odsetek, to fundusz PFR Inwestycje, możliwość podwyższenia kapitału. Tutaj jest nawet przewidziane 6 mld. To brak kar za opóźnienia w przetargach publicznych, to wreszcie przesunięcie utworzenia pracowniczych planów kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach na 1 października 2020 r. i szereg innych ułatwień, które zwalniają z biurokratycznych zadań. Wszystko to jest też po to, by właśnie chronić pracowników, by chronić miejsca pracy. To są rozwiązania przewidziane także dla rolników, o których nie zapominamy. To zatrzymanie windowania cen, które nieraz się dzisiaj odbywa. To świadczenie na dziecko w wieku do 8 lat. Szanowni Państwo! To jest nasz pierwszy, a nie ostatni krok. Kończąc pracę nad gospodarczą tarczą antykryzysową, nad tym pakietem, który tutaj przedstawiliśmy, rozpoczęliśmy jednocześnie prace nad kolejnymi ustawami, bo mamy kolejne takie pomysły, które mają ułatwić nam wyjście z tej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Myślę, że dzięki temu wysiłkowi, który podjęła pani marszałek, polegającemu na tym, że Sejm będzie także mógł pracować zdalnie, będziemy mogli na bieżąco szybko reagować i odpowiadać na zapotrzebowania rynku. Szanowni Państwo! Byłoby sprawą nieuczciwą składanie takich gwarancji, że tarcza pokryje przedsiębiorcom wszystkie poniesione koszty. Byłoby nieuczciwe z naszej strony mówienie, że jesteśmy w stanie zagwarantować wszystkim utrzymanie dotychczasowych dochodów, ale uczciwe jest zapewnienie, że robimy wszystko, by chronić miejsca pracy, że robimy wszystko, by chronić majątek Polaków. Wysoka Izbo! Wielokrotnie już jako Polacy dawaliśmy radę wyjść nie z takich opresji. Warunek jest jeden: musimy działać razem. Musimy działać razem, musimy dzisiaj być wspólnotą. Nie tylko tutaj, w Sejmie, nie tylko jako klasa polityczna, ale przede wszystkim jako naród, jako synergia działań rządu, samorządu, biznesu, przedsiębiorców. Wysoka Izbo! Dziś nie jest czas na kłótnie, dziś nie jest czas na robienie sobie zabawnych selfie, dziś nie jest czas na przerzucanie się odpowiedzialnością, dziś nie jest czas nawet na wzajemne obrzucanie się różnymi epitetami. Dziś jest czas na wspólną pracę dla Polski i do tej wspólnej pracy chcemy państwa gorąco zachęcać, bowiem w takich momentach, w momentach najbardziej dramatycznych, możemy rzeczywiście także zbudować coś wielkiego. Wyobraźcie sobie państwo - to jest historia autentyczna - kraj, który musiał się zmagać nie z takim kryzysem, a z tym, że poniósł cztery wielkie klęski, że stracił. My mówimy tutaj o tym, jak każde życie ludzkie jest cenne, że za każdym z nich kryją się nie cyfry, które są pokazywane, liczby zakażonych i zabitych, ale ludzkie dramaty i zawiedzione ludzkie marzenia.

Choć z innych powodów, bo nasi koledzy nie byli w sali obok, ale po prostu albo ich synowie nie żyli, albo oni nie żyli. Wyobraźcie sobie, że ten kraj był rzucony na kolana, ten kraj zbankrutował tak naprawdę, jak powiedział też pan premier o innych. Wtedy pomocy udzielili mu przedsiębiorcy, którzy dali kredyt państwu. Prosimy o wsparcie i ratowanie miejsc pracy. To były Ticinus, Trebia, Jezioro Trazymeńskie i Kanny. Tym państwem był Rzym, rzucony na kolana przez Hannibala. Po 14 latach odniósł druzgoczące zwycięstwo, a ci przedsiębiorcy, którzy pomogli, także byli w stanie odbudować swoje majątki. Wysoka Izbo! My nie żyjemy w tak dramatycznych czasach, my nie stoimy przed tak trudnymi problemami i tak wielkimi tragediami. Ale dziś, będąc razem (Dzwonek), możemy przypomnieć sobie wspólnie słowa Cypriana Kamila Norwida, że ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek.

Do tej pory tego nie było ze względu na podłączenie tego systemu, ale będziecie państwo widzieli mijający czas na mównicy. Proszę. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Jesteśmy tutaj od wczoraj. Jesteśmy tutaj od wczoraj w poczuciu odpowiedzialności, ale również w poczuciu tego, że ciąży na nas wielki obowiązek pomocy wszystkim, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Dzisiaj mówimy nie tylko o polskiej gospodarce i zdrowiu, ale również o wartościach, które nam wszystkim powinny przyświecać. Solidarność, wspólnota, poczucie zbiorowej odpowiedzialności to coś, co powinno dzisiaj mieć największą wartość. Ubolewam nad tym, że po raz kolejny państwo próbujecie dzielić Polaków. Ubolewam nad tym, że wbrew wielu apelom, które dzisiaj się pojawiają, dzielicie polskich pracowników na lepszych i gorszych, dzielicie polskich pracodawców na lepszych i gorszych, chcecie pomagać tylko wybranym, nie patrząc na to, że nie ma dziś znaczenia, czy pracownik pracuje w malutkim sklepie zatrudniającym trzy osoby, czy też w fabryce, w której zatrudnionych jest kilkaset osób, bo dokładnie tak samo te osoby będą dotknięte skutkami kryzysu. Dzisiaj po raz kolejny wykorzystujecie wielką światową tragedię do tego, by atakować wartości, na których budowana jest Wspólnota Europejska. To nie przystoi, panie premierze, by odwoływać się do doświadczeń II wojny światowej i jednocześnie wykazywać słabość Unii Europejskiej. Nie, panie premierze, to właśnie dzięki Wspólnotom Europejskim po II wojnie światowej udało się odbudować Europę, udało się zagwarantować pokój. I dzisiaj jak nigdy potrzebujemy również solidarności europejskiej, a nie ataku na wspólne wartości. Pan nie rozumie współczesnego świata, panie premierze. Pan nie rozumie tego, że wspólnota to nie tylko wspólnota waszej partii, [[Oklaski]] że wspólnota i odpowiedzialność są potrzebne właśnie w takiej chwili. Apelowaliśmy i prosiliśmy: przyjmijmy ten pakiet w zgodzie, ale również w poczuciu wielkiej odpowiedzialności. Pan mówi dzisiaj o tym, że każdy dzień to wielkie zagrożenie. Dokładnie tak. I wczoraj zajmowaliście się samymi sobą, zamiast przyjąć dobre rozwiązania. My dzisiaj składamy konkretne propozycje i konkretne poprawki. Chcemy, by rodzice, którzy dzisiaj są w domach, którzy dzisiaj otrzymują świadczenie, mogli otrzymywać je również po poniedziałku, kiedy wasze świadczenie się kończy, ale chcemy, żeby to świadczenie dostawali również opiekunowie osób z niepełnosprawnościami powyżej 8. roku życia i inni opiekunowie dzieciaków powyżej 8. roku życia. I prosimy, żebyście to rozwiązanie przyjęli. Prosimy również o to, byście nie dzielili przedsiębiorców na lepszych i gorszych, pracowników na lepszych i gorszych. Proponujemy odbiurokratyzowanie tego systemu, proponujemy czyste zasady dla wszystkich. O to błagają polscy przedsiębiorcy, ale o to błagają też polscy pracownicy. Proszę zrozumieć, że jeżeli uzależnicie pomoc państwa od przychodu, to dzisiaj pani, która prowadzi sklepik spożywczy, ma te przychody powyżej 15 tys. zł, tylko że dochodu nie ma żadnego, bo koszty stałe są większe. Dzisiaj pracodawca, który zatrudnia 11 osób w zamkniętej restauracji, będzie musiał zwolnić te osoby, bo wy wymyśliliście, że to ma być kryterium do 9 osób. Raz jeszcze apeluję: nie dzielcie Polaków na lepszych i gorszych. Dzisiaj jest wielki czas próby, dzisiaj jest czas próby dla nas wszystkich, by w poczuciu odpowiedzialności upomnieć się o elementarne zasady: solidarność społeczną, równość wobec prawa, ale również wspólnotę, która musimy razem odbudować. Dzisiaj do pakietu antykryzysowego staraliście się dopisać rozwiązania, które z walką z kryzysem nie mają nic wspólnego. Chcieliście, by prokuratorzy mogli ludzi zamykać w ich domach na 3 miesiące bez żadnej kontroli. To były wasze pomysły.

Proponujecie wyrzucić przestępstwo urzędnicze polegające na niedopełnieniu obowiązków lub przekroczeniu uprawnień. To jest wstyd, panie premierze, nigdy nie powinniście tego robić. Wreszcie, panie premierze, proszę się zastanowić, proszę raz jeszcze przemyśleć tę waszą strategię. Chcemy, byśmy ponad podziałami upomnieli się o tych wszystkich, którzy dzisiaj boją się o utratę miejsc pracy. Nie wprowadzajcie zapisów biurokratycznych, nie wprowadzajcie kategorii pracodawców i pracowników, nie wprowadzajcie pojęcia przychodu, kiedy ludzie nawet nie mają dochodu.

Bo pan, panie premierze, dziś jest premierem rządu Rzeczypospolitej, a nie prezesem banku. Odpowiedzialny szef rządu już dawno wprowadziłby stan klęski żywiołowej. Wiecie dlaczego? Właśnie dlatego, że dzięki takiemu stanowi klęski żywiołowej wy, polscy przedsiębiorcy, wy, którzy ciężko pracujecie na to, by budżet miał podatki, moglibyście starać się o odszkodowania.

Dzisiaj, wsłuchując się w głos pana szefa, bardzo zły, który mówi tylko i wyłącznie o interesie wyborczym, nie wprowadza pan stanu nadzwyczajnego. Bardzo dziękuję. Pani poseł. Chcę jeszcze tylko państwa poinformować, że w międzyczasie wpłynął wniosek naszego klubu o przejście do drugiego czytania bez odsyłania do komisji. Bardzo proszę, pani poseł. Wysoki Sejmie! Dzisiaj wszyscy jesteśmy na wojnie. Ale, panie premierze, pan nie jest wojnie z Unią Europejską ani z Koalicją Obywatelską, dzisiaj wszyscy jesteśmy na wojnie z wirusem, który niszczy zdrowie i życie Polaków i który niszczy zdrowie i życie polskiej gospodarki. Naszą odpowiedzialnością, odpowiedzialnością polityków jest dzisiaj ratowanie zdrowia i życia Polaków, zdrowia i życia polskiej gospodarki. Co trzeba zrobić dla systemu ochrony zdrowia, powie pani marszałek Kidawa-Błońska, bo apeluje o to od wielu tygodni. Ale co trzeba zrobić, aby wygrać wojnę o polską gospodarkę, o przyszłość Polski, żeby uratować miejsca pracy i firmy? Jak epidemiolodzy mówią: testy, testy, testy, tak ekonomiści mówią: płynność, płynność, płynność. Dzisiaj tej płynności dramatycznie potrzebują sklepikarze, fryzjerzy, kosmetyczki, ale równie dramatycznie potrzebują jej firmy, które zatrudniają 10, 15 czy 40 osób. Równie dramatycznie potrzebują firmy, które zatrudniają 100 i 1000 pracowników. Oni wszyscy mogą stracić pracę i zostać bez środków do życia. Reszcie to wirus powiedział: stop, dlatego musicie pokazać: stop należnościom dla fiskusa, dla ZUS-u od wszystkich firm, od wszystkich pracodawców i pracowników, którzy są dotknięci tą epidemią. Musicie także dać minimalne wynagrodzenie wszystkim pracownikom, nie 40%, nie w zależności od tego, czy firma straciła mniej czy więcej. Dzisiaj wszystkie firmy dotknięte epidemią muszą mieć pewność, że utrzymają miejsca pracy, ale tylko wtedy, jak na czas epidemii rząd pokryje z budżetu minimalne wynagrodzenie, bo ludzie nie dostaną pieniędzy od swojego pracodawcy. Jak chcecie zatrzymać ludzi w domu? Nie zatrzymacie głodnego człowieka w domu, on pójdzie, wyjdzie z domu szukać pieniędzy, żeby kupić jedzenie. Jeśli chcemy zatrzymać epidemię, o co apeluje minister Szumowski, to musimy ludziom zapewnić środki do życia na ten krótki czas. Musicie zaufać przedsiębiorcom. Nie możecie ich dzisiaj obarczać biurokracją. To musi być oświadczenie, przedsiębiorca składa oświadczenie. Jeśli nas nie posłuchacie, nie uratujecie ani firm, ani miejsc pracy, ani gospodarki.

Nie chcę, żeby pan mówił o 200 mld pomocy w czasie, gdy daje pan z budżetu państwa w 2020 r. na walkę z epidemią i jej skutkami 10 mld z budżetu państwa. Dzisiaj nie jest czas na oszczędzanie. Na to był czas przez 4 lata. Dzisiaj mówimy wam, my, liberałowie gospodarczy, że dzisiaj jest czas na wydawanie publicznych pieniędzy, żeby ratować zdrowie i życie ludzi, zdrowie i życie polskiej gospodarki. Nie wystarczy pomóc niektórym, nie wystarczy pomóc tylko trochę. Mówimy wam jeszcze raz: ludziom potrzebne są publiczne pieniądze bez propagandy, bez helikoptera.

Dziękuję. Bardzo proszę. Mówiłam wczoraj, że z koronawirusem nie wygra się kłamstwem. Wiem, że ta prawda jest bolesna, ale nawet najbardziej bolesna prawda pozwoli nam znaleźć dobre i mądre rozwiązanie. Nie pokonamy koronawirusa, jeżeli nie będziemy mieli zaufania. Ratownik medyczny musi mieć zaufanie do pacjenta, że powie mu prawdę, że jest zakażony. Pielęgniarka i lekarz muszą mieć zaufanie do ministra. Jeżeli on mówi, że jest sprzęt, że są medykamenty i są testy, to one naprawdę są. Widziałam dzisiaj wstrząsający materiał ratownika medycznego, który opowiadał, jak wygląda jego praca. Musimy mówić prawdę, nie możemy fałszować. Lekarz, dyrektor szpitala nie może zwalniać pielęgniarki tylko dlatego, że mówi prawdę. Nie może to mieć miejsca. My, panie ministrze, potrzebujemy, i wiemy o tym, więcej pieniędzy na ochronę zdrowia, na testy, na sprzęt, na środki ochrony, ale potrzebujemy także pieniędzy na to, żeby wesprzeć lekarzy i pielęgniarki, bo oni pracują bardzo ciężko. Muszą czuć, że państwo o nich w tym momencie dba.

Dlatego proponujemy, żeby z tych właśnie pieniędzy unijnych przeznaczyć 20 mld na stworzenie celowego funduszu właśnie na walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Bardzo pięknie jest na każdej konferencji wychodzić i mówić: dziękujemy wam za ciężką pracę, podziwiamy waszą misję, ale trzeba to docenić. Oni muszą teraz dostać nasze realne wsparcie. Możemy pomóc lekarzom także w inny sposób, pozwalając Polakom zostać w domu, o czym mówiła przed chwilą poseł Leszczyna. Jeżeli ludzie będą mieli zapewnione bezpieczeństwo ekonomiczne, zostaną w domu i łatwiej nam będzie opanować tę epidemię, ale musimy traktować wszystkich tak samo - i duże firmy, i małe, wszystkich pracodawców. Tutaj musimy być solidarni, nie możemy znowu dzielić Polaków. Dlatego jesteśmy gotowi do współpracy, bo ta tarcza, o której pan premier mówi, jest bardzo krucha i dziurawa. Wspólnie, jeżeli posłuchacie naszych rad, możemy z tego zrobić dobre narzędzie, żeby naprawdę Polacy czuli się bezpiecznie. Musicie także nas posłuchać, naszych rad, bo naprawdę wiemy, co mówimy. Dziękuję. Pan poseł Krzysztof Gawkowski, klub parlamentarny Lewica. Wysoka Izbo! Dziś jako społeczeństwo zdajemy egzamin z siły solidarności, z bycia wspólnotą, jaką państwo powinno być w tych trudnych chwilach. Być może jest to najpoważniejsza decyzja, jaką będziemy podejmowali w nadchodzących dziesięcioleciach. Najpoważniejsza próba, przed jaką stajemy w ciągu całego naszego życia. Wszyscy mierzymy się z epidemią, której skali nie jesteśmy w stanie oszacować. Znajdujemy się w przededniu wywołanego kryzysu gospodarczego, którego skutków również nikt nie jest w stanie przewidzieć. Ale wiemy jedno, że od naszych działań tu i teraz zależy, w jakiej kondycji będziemy po tym kryzysie. To od naszych decyzji podejmowanych niestety przy pustej sali zależy przyszłość milionów Polek i Polaków. Cały świat od 2 miesięcy toczy nierówną walkę z koronawirusem. To nie jest czas na to, żebyśmy na tej sali mówili o Rzymie, tylko o Polsce. To nie czas na polityczną walkę, to nie jest czas na zaczepki w Internecie i medialna nagonkę. Lewica nie będzie brała w tym udziału. Dziś liczy się tylko jedno. Polacy oczekują od nas, abyśmy szybko i sprawnie wprowadzili takie prawo, które pomoże ludziom bezpiecznie żyć, zabezpieczyć miliony Polek i Polaków. Lekarze, pielęgniarki, sprzedawcy, kasjerzy, listonosze, kurierzy, pracownicy magazynów, firm spedycyjnych, spółdzielcy, rolnicy, restauratorzy, służby mundurowe i wiele, wiele innych zawodów. Miliony z was pracują dzisiaj dzielnie, codziennie chodzą do pracy, ryzykują zakażenie wirusem, narażają siebie i swoje rodziny. Dziś dzięki ich poświęceniu nasze państwo i gospodarka funkcjonują. Z tego miejsca, z Sejmu, chciałbym wam wszystkim serdecznie podziękować. Nie zawiedziemy was. W tej Izbie mamy się spierać, bo po to ona jest. Jesteśmy po to, żeby dyskutować. Powinniśmy dzisiaj rozmawiać tylko o tym, jak pomóc polskim rodzinom, pracownikom, jak ratować gospodarkę i przedsiębiorców. To przesłanie przynosi dzisiaj do Sejmu Lewica. O to będziemy walczyli. Jeśli jednak mamy pracować, to bądźmy ze sobą szczerzy. Lewica nie będzie godzić się, kiedy premier zaklina rzeczywistość, że wszystko jest w naszym kraju w porządku. Powiedzmy sobie to uczciwie: można było zrobić więcej i lepiej przygotować się do epidemii. Rządzący przespali sporo czasu, kiedy wszystkie służby na świecie, polskie i zagraniczne, alarmowały. Zabrakło w magazynach maseczek, kombinezonów i płynów do dezynfekcji. Ale na rozliczenia przyjdzie czas, na konsekwencje również. W tym trudnym czasie powinniśmy być wspólnotą polityczną i społeczną. My jako Lewica taką współpracę deklarujemy. Musimy zrobić wszystko, żeby jak najszybciej wyjść z tego kryzysu. Proszę państwa, wczoraj liczba zakażonych przekroczyła 1000, dzisiaj wynosi ponad 1200. Choroba przyspiesza i my jako politycy również musimy przyspieszyć. Lewica była, jest i będzie blisko ludzi i codziennych ich problemów. Dziś rodacy potrzebują pomocy. Mają obawy, jak się utrzymać, czy dostaną pensje, czy zapłacą za czynsz, ratę kredytu czy za jedzenie.

Jesteśmy im to winni. Jako Lewica wielokrotnie deklarowaliśmy i dalej będziemy deklarować chęć współpracy. Nasz zespół ekspertów przygotował ponad 200 poprawek. Chęć współpracy nie oznacza, że będziemy bezkrytycznie przyjmować i popierać wszystkie propozycje rządu. Lewica ma obowiązek wobec obywateli, ale nie wobec władzy. Dlatego mówię jasno i wyraźnie: negatywnie oceniamy wiele propozycji rządowych. Widać w nich pośpiech, krótkowzroczność, czasem brak refleksji. Czasami są to rozwiązania zwyczajnie szkodliwe i niebezpieczne, antypracownicze i antyobywatelskie, za którymi Lewica nie podniesie ręki. Nie dopuścimy, aby aplikować dzisiaj lekarstwo, które może polskiej gospodarce zaszkodzić bardziej niż choroba. Nie dopuścimy, aby państwo przerzuciło koszty kryzysu na obywateli, pracowników i przedsiębiorców. Lewica nigdy się nie zgodzi, aby w ramach kryzysu rząd zafundował nam terapię szokową. W imieniu klubu Lewicy deklaruję jasno, że nie ma zgody na to, aby ukryć w przepisach obniżenie płac pracowników. Tym bardziej nie ma zgody na to, aby obniżyć pensje o połowę. Nie pozwolimy na ograniczenie odpoczynku i wydłużenie czasu pracy. Nie ma zgody na wprowadzenie tylnymi drzwiami ograniczeń praw i swobód obywatelskich. Nie ma zgody na to, aby ograniczać działalność organizacji pozarządowych. Nie zgadzamy się na wprowadzenie państwa do policyjnego aresztu, co dzisiaj chcecie nam zaproponować. 70% firm chce teraz zwolnić pracowników. Miliony ludzi wypchniętych na umowy śmieciowe lub samozatrudnienie już straciło pracę. Ci wszyscy ludzie potrzebują pomocy i wynagrodzenia. To nie są wykresy ani statystyki. To są ludzie, to są Polki i Polacy. To setki tysięcy rodzin pozostawionych bez środków do życia. Jeżeli interesuje was los tych wszystkich ludzi, to pamiętajcie, że z ich konsumpcji do tej pory żywił się budżet państwa. Jeżeli oni nie będą mieli pieniędzy, to nie wytłumaczymy tego tym wszystkim, którzy odpowiadają dzisiaj za politykę budżetową państwa. Ale gdzie są konkrety, panie premierze? Lewica kładzie je na stole i mówi wyraźnie: to jest nasz pakiet. Musimy rozszerzyć prawa pracownicze, żeby wszyscy mieli zagwarantowane wynagrodzenie, również ci, którzy są na samozatrudnieniu. Nie musimy dzisiaj mówić, że będziemy obcinali pensje. Dzięki temu pracodawca opłaci jedynie pozostałe 25% wynagrodzenia, ale tylko wtedy, kiedy utrzyma miejsce pracy. Musimy zagwarantować bezpieczeństwo milionów Polek i Polaków. Dziesiątki, setki tysięcy ludzi w Polsce patrzą w przyszłość z niepokojem. Wiedzą, że nie będzie ich stać na kredyty.

W czasach kryzysu musimy być solidni i solidarni, a nie żerować na nieszczęściu innych. Dlatego postulujemy również wprowadzenie i powołanie komitetu antyspekulacyjnego, który pozwoli, że nikt nie będzie hodował się na lichwie, że nie będzie nieuzasadnionych wzrostów cen. Oprócz pracowników, co mówimy jasno, są jeszcze przedsiębiorcy. Dlatego postulujemy, aby na czas kryzysu państwo przejęło finansowanie najmu, opłat leasingowych, energii elektrycznej i rachunków za gaz. Domagamy się również, aby pan premier wprowadził zwolnienie z płacenia przez naszych polskich przedsiębiorców podatku ZUS i innych podatków. Inaczej te firmy nie przetrwają. Jeśli milionom Polek i Polaków grozi dzisiaj bankructwo, to powinniśmy ich wspomagać. Cytował pan dzisiaj Stiglitza, ale ja rekomenduję, panie premierze, żeby czytać też jego wnioski. Nie odtworzymy gospodarki, jeśli zniszczymy dochody pracowników, obniżając im płace.

Nie wolno zakłamywać rzeczywistości o naszej europejskiej rodzinie. Dużym wsparciem jest Unia Europejska, która daje nam dzisiaj ponad 30 mld zł. Panie premierze, nie idźmy tą drogą. Na koniec ważna sprawa, która dotyczy ważnego sektora: opieki zdrowotnej. 7% nie wystarczy w obecnej skali pandemii na to, żebyśmy uchronili Polaków przed niebezpieczeństwem. Niecałe 8 mln zł w przeliczeniu na jeden szpital. Panie premierze, to zdecydowanie za mało. Potrzeby są ogromne. Z całej Polski docierają informacje, że brakuje zaopatrzenia. Dzisiaj rano rozmawiałem z jednym z dyrektorów szpitala w województwie kujawsko-pomorskim. Powiedział, że w tamtym tygodniu dzwonił kilkakrotnie do Ministerstwa Zdrowia. W tym tygodniu już nikt nie odbiera tam telefonów. Długo przed wybuchem epidemii Lewica biła na alarm w sprawie bankrutujących szpitali i zamykanych oddziałów. Ostrzegaliśmy, że to się źle skończy. Jeżeli premier Morawiecki znalazł 70 mld dla sektora bankowego, to tym bardziej powinien wiedzieć, że 7,5 mld na ochronę zdrowia wygląda marnie. Naprawdę priorytety są gdzie indziej. Z epidemią walczą nie tylko maseczki i rękawiczki. Z epidemią walczą ludzie: bohaterscy lekarze, pielęgniarki i cały personel medyczny. To przede wszystkim oni dzisiaj, i chylę przed nimi czoła, walczą jak bohaterowie z tą pandemią. I im należy się również rekompensata. Dlatego Lewica apeluje: przyjmijcie naszą poprawkę przewidującą dodatkowe 50% stawki dla pracowników szpitali.

Dziś jednak czas wesprzeć finansowo również lekarzy na pierwszej linii frontu. Szanowne Panie Posłanki i Panowie Posłowie! Na zakończenie zwracam się do was z apelem: proszę o wspólną, merytoryczną i spokojną pracę nad tą ustawą. Życie i zdrowie Polek i Polaków nie ma barw partyjnych. Epidemia nie ma sympatii politycznych. A jeśli chcemy skutecznie poradzić sobie z epidemią, musimy współpracować. Podobnie nie ma znaczenia to, z jakiej opcji przychodzimy, czy jesteśmy dzisiaj rządem, czy opozycją, czy poprawki są z Lewicy, PSL-u, Platformy, czy PiS-u. Te rozwiązania mają być dobre dla Polski. W obecnym kształcie tarcza antykryzysowa nie jest wystarczająca i pan premier wie to doskonale. Jest ona również czasami bardzo antyprzedsiębiorcza, szkodliwa, przeciwskuteczna - i to też trzeba sobie otwarcie powiedzieć. Jesteśmy gotowi do merytorycznej pracy przed ostatecznym uchwaleniem ustawy. Prezentował je nasz kandydat na prezydenta Robert Biedroń. Jeszcze raz apelujemy o to, co we wstępie. Zróbmy wszystko, żeby to posiedzenie nie trwało kilka godzin, żebyście walcem nie przejechali tej ustawy, żebyśmy mieli prawo pomóc pracowniczkom i pracownikom. Obywatele inaczej nam tego nie wybaczą, tego, że przyjmujemy złe prawo. Liczymy na odpowiedzialne zachowanie rządu. Lewica zrobi wszystko, aby w dobie kryzysu nikt nie został sam. Ani przedsiębiorcy, którzy w tej chwili walczą o zachowanie miejsc pracy, ani miliony pracowników, którzy dzisiaj nie są pewni nawet jutra. W tej chwili walczymy o to, żeby Polacy, 38 mln Polek i Polaków, mogli godnie żyć.

Mówimy głosem małych, mikro- i średnich przedsiębiorstw, których brak państwa pozbawi możliwości funkcjonowania i zbankrutują. Upominamy się o pracowników opieki zdrowotnej, która od lat cierpi na chroniczne niedofinansowanie. Mówimy głosem spółdzielców i rolników. Mówimy dzisiaj odpowiedzialnie. Jeżeli chcemy, żeby to prawo służyło Polkom i Polakom, wszyscy musimy się zjednoczyć. Ale nie możemy iść jak walec przez te ustawy tylko dlatego, że trzeba je przyjąć w ciągu 3 godzin. Lewica nie zgodzi się na to, żeby ograniczać prawa pracownicze milionów Polek i Polaków. Nie może być tak, że ci właśnie ludzie zapłacą za ten kryzys. To jest warunek Lewicy, jeśli chodzi o poparcie tego projektu. To jest ten mur, który budujemy. Albo Polki i Polacy zobaczą, że chcemy im pomagać, zobaczą, że w tej Izbie jest zgoda, zobaczą, że jesteśmy razem z nimi, albo nam nigdy tego nie wybaczą. To jest warunek Lewicy, z którego się nie wycofamy, bo nasza odpowiedzialność nie jest przed rządem, jest przed obywatelami i obywatelkami, jest przed naszymi rodakami, jest przed Polską. Lewica zawsze będzie po waszej stronie. Dziękuję bardzo.

Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - PSL - Kukiz15 chcę zabrać głos w jednej z najważniejszych debat ostatnich dziesięcioleci. Panie premierze, na początek taka prośba. Proszę uświadomić swoim ministrom, że nie biorą udziału w rekonstrukcji bitwy pod Kartaginą, tylko w walce z koronawirusem o miejsca pracy, o zdrowie i życie, o polską gospodarkę. To znaczy: trzeba zejść na ziemię. Nie jesteśmy na spotkaniu kółka historycznego, tylko w polskim parlamencie, i rozmawiamy o życiu i zdrowiu polskich pacjentów, polskiej gospodarki, o ratowaniu nas przed armagedonem gospodarczym. Ludzie, ogarnijcie się. Jak wy się zachowujecie? Naprawdę przyjdzie czas na dyskusje panelowe, historyczne. Najpierw trzeba postawić rozpoznanie. A rozpoznanie jest takie, że koronawirus zaatakował nas nie tylko biologicznie - są poszkodowani pacjenci, są całe rodziny, które są dzisiaj przerażone, są pracownicy ochrony zdrowia, którzy każdego dnia walczą o zdrowie i życie - ale także zaatakował polską gospodarkę. W najbliższych tygodniach może dojść do masowych zwolnień, zwolnień grupowych w wielu zakładach pracy. Co druga polska firma może upaść. Taka jest sytuacja i to jest dzisiaj postawione rozpoznanie i diagnoza. Jakie zastosować leczenie? Co zrobić, żeby uratować dzisiaj każde miejsce pracy? Tak jest, solidarność Polaków, zdajemy egzamin z solidarności, pomocy sąsiedzkiej, pomocy jeden drugiemu. Zdają egzamin z solidarności pracownicy ochrony zdrowia, bo pomimo braków w sprzęcie ochronnym są na pierwszej linii walki. Nie zabezpieczyliście ich. To jest zaniedbanie, z tego będziecie rozliczeni. Ale oni walczą i zdają egzamin z solidarności. I teraz jest pytanie do nas wszystkich tu, na tej sali, wszystkich parlamentarzystów: Czy my zdamy egzamin z solidarności? Czy jesteśmy gotowi przerwać te nasze wojenki, schować to wszystko, te uszczypliwości i normalnie zastosować zasadę solidarności? Ale solidarność musi być dwukierunkowa.

Bo jak mówiliśmy o dobrowolnym ZUS-ie 2 tygodnie temu, 2 miesiące temu, to był to dla was koncert życzeń, były to pobożne życzenia, ale jak podpisał się pod tym pan prezydent, to mówicie: tak, to jest dobry pomysł. Nie lansujcie Andrzeja Dudy, bo to i tak mu nie pomoże, a może zaszkodzić wielu polskim firmom, bo nie wiedzą, co się dzieje, bo te komunikaty po posiedzeniu Rady Gabinetowej były tak miałkie i tak beznadziejne, że kompletnie nic z tego nie wynikało. Druga sprawa. Jak opozycja dzisiaj zgłasza nawet trudne na pierwszy rzut oka do przyjęcia poprawki, to pochylcie się nad nimi. Dziękuję. To kompletnie nie ma sensu. Konkretne działanie. Dobrowolny ZUS, i to niezależnie od wielkości firmy, bo koronawirus nie działa punktowo, że atakuje tylko mikroprzedsiębiorstwa, on atakuje wszystkie. Zwolnienie z PIT-u, z CIT-u. Zwolnienie, a nie przełożenie. Tak samo w sprawie kredytów. Trzeba nie tylko zastosować wakacje kredytowe, ale też wydłużyć okres spłaty kredytu, bo ktoś może mieć kredyt do spłaty jeszcze przez 7 miesięcy, skorzysta z wakacji kredytowych przez 6 miesięcy. To jest kompletnie bez sensu. Nieoprocentowane pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego. O tym będzie mówił marszałek Tyszka. Nie 5 tys. z Funduszu Pracy. Pan premier mówił, jak to zachowaliście bezpieczne instrumenty, jak to zabezpieczyliście fundamenty finansowe. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Panie premierze, ile tam jest pieniędzy? A on ma starczyć na wypłaty. Ta wypłata wynagrodzeń musi być. Rozumiem wnioski Lewicy. Pamiętajcie, żeby też nie przeszarżować, ale rozumiem waszą walkę o prawa pracownicze. My mówimy wprost: minimalne wynagrodzenie dla każdego pracownika, którego firma ucierpiała. To naprawdę nie ma sensu. Tak nie pomożemy. Proste, jasne reguły. Bez oświadczeń i zaświadczeń na cztery, pięć stron.

Dla pana premiera, bo powoływał się na to, ważne są opinie ekspertów instytutów ekonomicznych. Panie premierze, dla mnie w czasie kryzysu ważna jest opinia prawdziwych ekspertów: polskich przedsiębiorców. Pani Hanny, która prowadzi biuro podróży, pana Stanisława, który ma firmę transportowa, i pana Jana, który napisał do mnie przed chwilą: trochę lipa, że rząd bierze pod uwagę przychód, a nie dochód, i to z lutego, np. ja mam małą marżę, ale przychód w lutym miałem ponad 15 600 i ZUS będę musiał zapłacić, mimo że w marcu już mam megaspadek przychodu, a dochodów prawie zero. To jest głos prawdziwego eksperta. Szukajcie tych ekspertów wśród polskich przedsiębiorców, polskich pracodawców. Dobrze, że dopisaliście rozwiązania dla rolników.

Ratujmy każde miejsce pracy. Upominam się również o polskie samorządy. Musi dojść do zwolnienia z podatku od nieruchomości, z podatku rolnego, do umorzenia tych podatków na najbliższe miesiące, musi być wsparcie dla samorządów ze strony rządu. Nie można zostawić małej wspólnoty lokalnej samej sobie. Oni już dzisiaj mają wielkie problemy choćby z utrzymaniem szkoły, z wypłacaniem wynagrodzeń dla nauczycieli. Po tym armagedonie gospodarczym mogą po prostu upadać. Tu chodzi też o spółki komunalne. Mamy do zrealizowania ogromne przedsięwzięcie przeprowadzenia Polski przez kryzys, jakiego nie znaliśmy, jakiego nie doświadczyliśmy. Stoimy nad przepaścią. Jedni są sparaliżowani strachem, nie wiedzą, jak się zachować, drudzy chcą iść na oślep, choćby bez oręża. Zasada solidarności, zasada pomocniczości, zasada odpowiedzialności jeden za drugiego. Nie można pozostawić lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów i farmaceutów samym sobie. Trzeba im zapłacić lepiej za ten czas bardzo wytężonej pracy.

Co mają zrobić pacjenci onkologiczni, po przeszczepach, z chorobami, którzy nie mogą czekać? Musicie ich o tym informować. My jesteśmy gotowi do współpracy, ja tę współpracę jeszcze raz deklaruję. Spełnijcie kolejne nasze postulaty zawarte w poprawkach: dobrowolny ZUS dla wszystkich, CIT, PIT zamrożony, niepobierany, szybki zwrot VAT-u, podatek od nieruchomości, wynagrodzenia dla pracowników w minimalnym... minimalne wynagrodzenie dla każdego pracownika, który tego wsparcia potrzebuje, zasiłki nie do 8. roku życia, tylko również na opiekę nad starszymi dziećmi. To są nie warunki, to są nasze żądania, powiem wprost. One są po prostu potrzebne, bo są żądaniami pracowników i pracodawców. Zróbmy to wspólnie. Jak najszybciej trzeba to prawo uchwalić, ale musi być mądrze uchwalone i dobrze uchwalone. Mam nadzieję, że są przygotowane akty wykonawcze, są przygotowane rozporządzenia, bo to musi być natychmiast. I na koniec wniosek do pana marszałka: Sejm nie powinien przerywać swoich obrad, powinien pracować w trybie ciągłym, każdego dnia. Każdego dnia ma się odbywać posiedzenie. Za 2 tygodnie oczekuję od pana premiera raportu na temat wdrożenia ustawy antykryzysowej.

Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Będę mówił mniej politycznie, a bardziej o gospodarce i o przedsiębiorcach. Światowa i polska gospodarki wyglądają w tym momencie jak człowiek postrzelony z armaty, natomiast nasz rząd na czele z panem premierem Morawieckim przychodzi z gencjaną i plasterkiem i w ten sposób chce uratować sytuację. To nawet nie jest ćwierćśrodek, to całkowicie odbiega od tego, co pan premier w swoim wystąpieniu na początku mówił, czyli że rzeczywiście mamy prawdopodobnie do czynienia z kryzysem największym od wielkiego kryzysu z przełomu lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Mamy do czynienia z sytuacją absolutnie bez precedensu, która wymaga natychmiastowego wdrożenia radykalnych działań. Wiedzą to najpotężniejsze państwa świata, takie jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja czy Niemcy. Rządy i banki centralne tych państw wprowadzają olbrzymie, szeroko zakrojone programy pomocowe na skalę dużo większą niż wprowadza Polska. Niestety mówię to z przykrością, dlatego że cenię ten gest w postaci ostatnich konsultacji. Natomiast cały czas mamy sytuację, w której prezes Narodowego Banku Polskiego pan Glapiński jeszcze parę dni temu mówił, że będziemy mieli w tym roku wzrost PKB o 2%. No to są oczywiście bajki, dlatego że za chwilę możemy mieć sytuację, w której upadną setki tysięcy polskich firm, miliony ludzi stracą pracę, jeżeli nie zostaną podjęte natychmiast radykalne, dużo bardziej radykalne działania. Mam wrażenie, że tę tarczę napisali urzędnicy na potrzeby urzędników. Zamiast prostych, automatycznych mechanizmów tarcza zakłada skomplikowane biurokratyczne procedury, składanie wniosków z dziesiątkami załączników i zabezpieczeń dla biurokratów. W ten sposób, szanowni państwo, będziemy mieli megarecesję i nigdy z tego nie wyjdziemy. My przeprowadziliśmy jako Kukiz15 bardzo szybkie konsultacje z naszym bezpośrednim zapleczem, czyli z tysiącami przedsiębiorców, dostaliśmy w ciągu paru godzin chyba ponad 1 tys. maili i wyciągnęliśmy z nich 10 postulatów, które wysłaliśmy do pana premiera. Teraz pozwolę sobie je odczytać, dlatego że one są zaskakująco powtarzalne. Po drugie, wprowadzenie powszechnej abolicji dla firm od danin publicznoprawnych, przede wszystkim PIT, CIT, VAT oraz składki na ZUS na 3 miesiące. Odroczenie terminów złożenia sprawozdań i deklaracji podatkowych co najmniej do 1 lipca. Wakacje kredytowe i leasingowe na 3 miesiące plus kolejne 3 miesiące odroczenie spłaty rat. Kwota wolna od podatku PIT dla wszystkich - 30 tys. zł. Odroczenie bądź obniżenie opłat za najem, czynsz na czas epidemii oraz zwolnienie z podatku od nieruchomości wraz z rekompensatą dla samorządów. Zwiększenie limitu nieoprocentowanych pożyczek do 50 tys. zł dla mikro-, małych i średnich firm. Możliwość odliczenia dla przedsiębiorców straty z 2020 r. od dochodu z 2019 r. Wypłata zasiłku chorobowego od pierwszego dnia przestojowego. Szanowni Państwo! Niektóre z tych postulatów zostały częściowo spełnione. To absolutnie nie wystarcza, żeby powstrzymać w tym momencie upadek setek tysięcy polskich firm. Cenię wrażliwość społeczną lewicy, natomiast to jest tak, że jeżeli będziemy myśleć tylko w kategoriach pracowników w tym momencie, to ci pracownicy nie będą mieli dokąd wracać. Przede wszystkim musimy uratować setki tysięcy polskich firm. Przypomnę, że mamy w Polsce 2 mln polskich firm, które zatrudniają 10 mln osób.

Słyszałem z ust przedstawicielki Platformy Obywatelskiej o tym, że przedsiębiorcy mówią: płynność, płynność, płynność. To prawda, mi też wszyscy przedsiębiorcy, z którymi rozmawialiśmy, to powtarzali, natomiast my chcieliśmy przedstawić konkretny projekt tego. Został wysłany do pani minister Emilewicz, chętnie opublikujemy to publicznie. Fundusz płynności - złożyliśmy już tę poprawkę do tej ustawy - z którego mają być finansowane opłaty za najem oraz wszystkie zobowiązania o charakterze ciągłym wszystkich przedsiębiorców. Fundusz będzie obsługiwał Bank Gospodarstwa Krajowego, a wnioski będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 3 dni przy minimalnych formalnościach. Wszystko będzie można załatwić elektronicznie i bez konieczności przesyłania tysięcy papierków. Wzorem niemieckim fundusz nie będzie miał górnego limitu (Dzwonek) i będzie dostępny dla wszystkich firm bez względu na wielkość. Dokładnie tego chcą polscy przedsiębiorcy. Bardzo proszę państwa, wsłuchajcie się w ich głos. Przeczytajcie choćby, panie premierze, apel branży meblarskiej zatrudniającej blisko 200 tys. osób. To jest coś.

Ja sobie zdaję z tego sprawę, że to jest niekonwencjonalne doprowadzić do dużego zadłużenia państwa, ale jesteśmy na etapie, w którym wszystkie państwa będą się zadłużały.

Panie Marszałku! Panie Premierze! Doczekaliśmy się tego momentu, w którym możemy dyskutować wreszcie o tarczy antykryzysowej. Po wielu dniach, po wielu tygodniach zapowiedzi, w czasie, kiedy inne rządy uruchomiły już proste rozwiązania dające wsparcie lub ujmujące ciężarów przedsiębiorcom, możemy dyskutować. Możemy dyskutować nad rozwiązaniami, które zaczną działać być może za miesiąc, być może za kwartał, a być może nie wiadomo kiedy, ponieważ wprowadzacie państwo w swoich propozycjach 24 nowe procedury administracyjne, które w tej chwili jeszcze nie istnieją, w momencie kiedy wiele urzędów przeszło na pracę zdalną albo jest sparaliżowanych, podobnie jak wiele firm w Polsce. Panie Premierze! Już w tej chwili tysiące osób zostały zwolnione. W poniedziałek i wtorek, ostatnie dni tego miesiąca, kolejne osoby dostaną wypowiedzenia. Zaproponowane przez was rozwiązania na rzecz rynku pracy zaczną działać za wiele miesięcy. To jest narzędzie całkowicie niedopasowane do potrzeb. Są cztery proste sposoby, które powinny być wykorzystane w tarczy antykryzysowej, którą powinien zaproponować rząd. Pierwsze - utrzymanie wynagrodzeń natychmiast, tu i teraz, dla firm, które nie mogą działać. Drugie - zwolnienie z ZUS i podatków. Jeżeli jest kwota pieniędzy, którą rząd chce przeznaczyć na pomoc, cała ta kwota powinna zostać podzielona pomiędzy działające przedsiębiorstwa i powinno się im umożliwić zwolnienie automatyczne, bez pisania żadnych wniosków - najprostsza procedura na świecie. Trzecie - dostęp do kapitału obrotowego bez żadnych specjalnych procedur, preferencyjny kredyt. Czwarte i ostatnie - wycofanie wszelkich nowych podatków. Pani minister Emilewicz obiecywała, że podatek cukrowy nie wejdzie. W tej chwili słyszymy, że te zapowiedzi są nieaktualne. Niestety te cztery proste rozwiązania nie są w obszarze zainteresowania rządu. Zamiast tego mamy całą paletę rozwiązań niezwykle skomplikowanych, których wprowadzanie i wdrażanie zajmie wiele miesięcy. Niektóre z zapowiedzi sformułowanych przez pana premiera zaczną działać za rok albo za 2 lata, jak np. inwestycje infrastrukturalne, których kwota została wliczona do tych 200 mld, czysto medialnych. Jesteśmy po tygodniu teatralnych konsultacji. W poniedziałek na spotkaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego nikt nie znał projektów rządowych, a mieliśmy wszyscy udawać, że nad nimi dyskutujemy. Dlaczego jesteśmy wciągani w takie teatralne konsultacje? To dziś, bo projekty ustaw są znane od wczoraj w nocy, zaczęła się realna dyskusja. Ale państwo chcecie wszystko dziś przegłosować. Czyli nasz głos, głos społeczeństwa, głos organizacji gospodarczych, tak naprawdę nie ma znaczenia. Jesteśmy tu tylko po to, żeby to przegłosować. Dobrze, zrobimy to. Przygotowaliśmy 39 poprawek, które za chwilę złożymy. Spróbuję szybko omówić główne kierunki, w których chcemy iść, próbując udoskonalić to, co przyniósł rząd. Pierwsza sprawa spośród tych 19, które wymienię: zwolnienie z ZUS dla wszystkich przedsiębiorców z mocy prawa, nie tylko dla niektórych i nie na wniosek. Tyle, ile nas stać, panie premierze. Tyle, ile chcecie zwiększyć deficyt budżetowy, o czym przed chwilą była mowa. Drugie - umorzenie ZUS dla najbardziej dotkniętych kryzysem branż i z mocy prawa, a nie tylko dla niektórych firm i na wniosek.

Złożymy w tej sprawie poprawkę. Czwarte - uwolnienie środków zamrożonych na rachunkach split payment. Piąte - dopłaty do wynagrodzeń natychmiast i przez 6 miesięcy, a nie po biurokratycznej ścieżce zdrowia i przez 3 miesiące. Szóste - wynagrodzenie postojowe w wysokości minimalnej krajowej w całości płacone przez państwo, a nie częściowo płacone przez pozbawionego dochodów pracodawcę. Siódme - dopłaty do wynagrodzeń i postojowe bez obowiązku utrzymywania miejsca pracy po zakończeniu kryzysu. Usztywnianie działania przedsiębiorstw w czasie kryzysu nie może dać dobrego efektu, bo przedsiębiorcy muszą adaptować się do zmieniających się okoliczności gospodarczych. Oczekiwanie, że w tej chwili pracodawcy zawrą swego rodzaju kontrakt z rządem, że nikogo nie zwolnią, po to, żeby dostać jakąś pomoc, jest działaniem zupełnie przeciwskutecznym. Racjonalny przedsiębiorca nie zdecyduje się na to. To jest nieracjonalne. To powiedziałem. Ósme - wypłaty zasiłków chorobowych z ZUS od pierwszego dnia. To też sposób na to, jak ulżyć przedsiębiorcom w kosztach stałych. Nie trzeba stworzyć żadnych komisji urzędniczych, żeby wprowadzić tę ulgę. Po prostu trzeba zmienić przepis. Dziewiąte - odroczenie do 30 września wszystkich deklaracji obowiązków sprawozdawczych, a nie tylko niektórych i tylko do czerwca. Panie premierze, w tym tygodniu zaczepił mnie przedsiębiorca, kiedy wchodziłem do swojego banku, i spytał: Dlaczego ministerstwo zapowiada wydłużenie sobie czasu na interpretacje podatkowe, i to o miesiące, a nie odsuwa czasu złożenia deklaracji podatkowych? To jest działanie totalnie antybiznesowe. Kredyty i leasingi to jedna z głównych pozycji w kosztach stałych przedsiębiorstw. Jedenaste - ustawowe zawieszenie spłat kredytów i pożyczek dla pracowników objętych przestojem oraz osób pobierających wsparcie dla samozatrudnionych i zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Dwunasta nasza propozycja - dopłaty budżetowe do kosztów lokali przedsiębiorców objętych spadkiem obrotów lub przestojem. Tu drobna uwaga. Konstytucjonaliści już podnoszą, że niewprowadzenie nadzwyczajnego stanu jest, po pierwsze, deliktem konstytucyjnym. I jednocześnie unikacie rekompensaty strat majątkowych, wynikającej ze specjalnej ustawy. Gdyby był stan nadzwyczajny, rząd miałby ten obowiązek. Nie wprowadzając stanu nadzwyczajnego, rząd ten obowiązek z siebie zdjął. To jest delikt konstytucyjny. Następna sprawa - wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju dla polskich przedsiębiorstw, a nie dla zagranicznych spółek. Tu złożymy również poprawkę.

Mianowicie, dopłata do pensji oraz zwolnienie z ZUS, a nie tylko jedno do wyboru. Składamy poprawkę - liczymy, że zostanie ona uwzględniona - aby można było korzystać jednocześnie z dopłat do pensji i ze zwolnienia z ZUS, a nie żeby przedsiębiorca musiał wybierać. Piętnaste - sprzeciw wobec wykorzystywania tarczy antykryzysowej do powiększania ucisku fiskalnego i uprawnień ZUS. Wczoraj pani minister Emilewicz przyznała się, że ewidencjonowanie przez ZUS umów o dzieło jest wstępem do tego, żeby je ozusować. Szesnaste - nie zdejmować odpowiedzialności z urzędników. Siedemnaste - epidemia nie może być pretekstem dla zwiększania władzy prokuratury. Wprowadzanie w tej chwili aresztów domowych to jest jakieś kompletne nieporozumienie. Osiemnasta sprawa. Metoda kasowa rozliczania VAT, którą proponujemy, żeby ulżyć przedsiębiorcom. Jak można zaproponować nieograniczone ceny maksymalne? Dwudziesta sprawa - tarcza biurokratyczna. 24 nowe wnioski i procedury. Tu są nasze poprawki. Proponujemy je. To dwie poprawki do ustawy o systemie ochrony zdrowia - będziemy za chwilę je składać - aż 32 poprawki do ustawy głównej antykryzysowej i pięć poprawek do ustawy o funduszu rozwoju. Dostaliśmy dzisiaj zaledwie 23 minuty na omówienie tego wszystkiego. To są poprawki merytoryczne. Nasi eksperci, nasi prawnicy pracowali nocami, ponieważ nocami zostały nam te projekty dostarczone. Mimo to dla dobra obywateli, dla dobra polskich przedsiębiorców nie odrzucamy tej szansy. Bardzo prosimy, proszę przyjrzeć się tym poprawkom, proszę z nich skorzystać. Proszę nie tworzyć nowych procedur urzędniczych, tylko wprowadzić automatyzm. Pan poseł Jakub Kulesza, koło Konfederacji. Wysoka Izbo! Mam wrażenie, że państwo nie zdają sobie sprawy z powagi sytuacji, w jakiej znaleźli się pracodawcy i pracownicy. Do dzisiaj pracodawcy wstrzymują się z decyzjami w nadziei na rozwiązania, które już funkcjonują w innych krajach, wstrzymują się z decyzjami, czy ciąć wydatki, czy zamykać przedsiębiorstwo, czy zwalniać ludzi. Dzisiaj rozstrzyga się przyszłość milionów polskich rodzin. Jak to zrobić, żeby pokazać, że się pomaga wszystkim, ale żeby nikomu nie pomóc? Niestety to tarcza biurokratyczna. Wszystkie te aspekty, o których przed chwilą mówił Krzysztof Bosak, sprawiają, że pracodawca teraz stanie przed ogromnym dylematem. Po pierwsze, czy ma skorzystać z ulgi na swój ZUS, czy skorzystać z dopłaty do podstawowego pracownika. Po drugie, czy podjąć ryzyko - bo on nie wie, co będzie za miesiąc, 2, 3, 4 miesiące - i skorzystać z dopłat do pracownika, ale będzie miał obowiązek utrzymania tego pracownika. To wszystko kieruje się w stronę takiego rozwiązania, że pracodawca powie: dziękuję, zamykam interes. To nie są rozwiązania, które pomogą utrzymać miejsca pracy w Polsce. Niestety, te rozwiązania mają służyć, mam wrażenie, tylko urzędnikom. Wprowadzanie ewidencji, ozusowania umów o dzieło w momencie i w sytuacji kryzysu jest całkowicie absurdalne.

Państwo powinni w takiej sytuacji wysłać też do kwarantanny podatki i opłaty, ponieważ nie będzie z czego ich opłacać. Szanowni Państwo! Wnoszę o to, by jak najszybciej wdrożyć poprawki przedstawione przez Konfederację, bo tylko to zapewni jak najszybsze wsparcie miejsc pracy tak, by Polacy mieli za co jutro kupić chleb. Dziękuję bardzo. Teraz połączymy się zdalnie z panem Konradem Berkowiczem z sali, w której on przebywa. Bardzo proszę o połączenie. Panie Marszałku! Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać, bo to pierwsze w historii Sejmu takie wystąpienie on-line. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać, bo to są rzeczy poważne. Polscy przedsiębiorcy w efekcie pandemii, w efekcie działań rządu stoją w obliczu rychłego bankructwa. Polscy przedsiębiorcy musieli przestać działać, nie mogą zarabiać, a nadal muszą płacić haracz w postaci rozmaitych podatków i składek ZUS dla państwa. Tymczasem tarcza antykryzysowa jest skonstruowana tak, żeby niemal nikt nie mógł z niej skorzystać, żeby niemal nikt nie mógł skorzystać z rozmaitych ulg podatkowych. Ona skreśla przedsiębiorców brutalnie, a reszcie Polaków mydli oczy, że rząd robi coś z gospodarką. Dlatego z całą mocą apeluję do pana premiera Morawieckiego, żeby zrealizował, poza pozostałymi poprawkami dziś przedstawionymi przez moich kolegów, m.in. postulat Konfederacji jeszcze z wyborów parlamentarnych i zwolnił przedsiębiorców i pracowników z obowiązku płacenia ZUS-u przynajmniej na czas tego kryzysu, bo nas nie stać teraz, żeby topić pieniądze w tej czarnej dziurze, jakim jest ZUS. To, że przedsiębiorcy obecnie noszą czasem maski na twarzach, nie oznacza, że można pluć im w twarz, a tym jest ta tzw. tarcza antykryzysowa. Pan poseł Grzegorz Braun, również zdalnie z sali 102. Bardzo proszę. Czy mamy połączenie z panem posłem?

Chciałbym zauważyć, że czas mojego wystąpienia biegł, jeszcze zanim miałem okazję je zacząć. To taki drobiazg, groteska, w jaką obróciliście obrady Wysokiej Izby. Obywatele to widzą, nasi rodacy. Tutaj nie ma miejsca i nie ma czasu na to, żeby poważnie rozmawiać nie o kryzysie, tylko o rezultacie tych działań, które podjęła administracja centralna warszawska pod pretekstem nie w pełni rozpoznanego zjawiska, które jedni określają jako akt wojny biologicznej, a inni decydują się wierzyć temu, co donoszą światowe mass media. Te światowe mass media ani też warszawskie nie tłumaczą, dlaczego np. już przed tygodniem ten słynny wirus o numerze 19 spadł z brytyjskiej listy chorób definiowanych jako szczególnie ryzykowne - high consequence infectious diseases. Jest taka strona rządu brytyjskiego i oni właśnie zmienili kategorię tego wirusa, co nie zmienia rzecz jasna linii postępowania rządu warszawskiego, którego - jasna rzecz - brytyjskie rozstrzygnięcia nie obowiązują, ale jednak idąc za przykładem z zagranicy, rząd warszawski jak za panią matką schładza do temperatury zerowej polską gospodarkę. I tu nie będzie okazji do tego, żeby się upomnieć w tych wszystkich sprawach, w których Konfederacja składa poprawki.

Dziękuję. Bardzo proszę. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zgłaszam wniosek o skierowanie projektów ustaw do komisji: Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Zdrowia.

Dziękuję. Lista zgłoszonych. Zgłosiło się do pytań pięć osób. Zamykam listę zgłoszonych. Bardzo proszę, pani poseł Maria Janyska.

Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! 2 tygodnie temu pan premier zapowiedział, że będziemy mieli najlepszy na świecie pakiet antykryzysowy. I przez te 2 tygodnie świat gospodarki: przedsiębiorcy mali, mikro, średni, duzi, pracownicy, zleceniobiorcy itd., itd. czekali z nadzieją na rozwiązania i zadawali sobie w tym czasie pytanie, co będzie jutro. Zadawali sobie to pytanie, bo wielu z nich już nie miało pracy w tym czasie, wielu z nich już zaprzestało działalności gospodarczej, a dla wielu z nich ten dzień miał nadejść lada moment. Wczoraj ukazał się ostateczny projekt. I jakie pytania dzisiaj zadają te grupy? I tych pytań: dlaczego, jest mnóstwo. Dlaczego te rozwiązania nie są powszechnie adresowane do wszystkich, których dotyka ten kryzys? Dlaczego powszechnie nie są anulowane daniny publiczne na czas kryzysu bez zbędnej biurokracji, tylko na oświadczenia. Dlaczego wszyscy nie mogą skorzystać z anulowania składki ZUS-u, podatków: PIT-u, CIT-u, dlaczego wszyscy nie mogą mieć zagwarantowanych najniższych wynagrodzeń na czas kryzysu, żeby można było przetrwać i to uratować? Dlaczego ta tarcza na samym wstępie już nie starcza? I teraz wszyscy, którzy siedzicie przy tabletach, członkowie komisji gospodarki, Zjednoczonej Prawicy weźcie sobie to do serca, weźcie te wszystkie pytania, które macie, do serca, zagłosujcie za poprawkami Koalicji Obywatelskiej (Dzwonek), która odpowiada na te pytania i podaje rozwiązania. Pan poseł Dariusz Wieczorek, klub Lewicy.

Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Rzeczywiście, tak jak przewodniczący Gawkowski mówił, 70% firm obecnie chce zwalniać swoich pracowników i zastanawia się nad zwolnieniami, nad obniżeniem pensji. W związku z tym mam pytanie do pani minister, czy rząd rzeczywiście analizuje sytuację na rynku pracy i szacuje, jaką potencjalnie grupę pracowników mogą objąć te restrykcje wynikające z aktualnej sytuacji. Kolejne pytanie: Czy rząd planuje, jeżeli chodzi o urzędy pracy, wsparcie urzędów pracy? Bo należy się spodziewać, że mimo wprowadzania tych ustaw, mimo tych działań osłonowych, liczba bezrobotnych na rynku jednak wzrośnie, a to spowoduje, że te urzędy pracy będą miały zdecydowanie więcej zadań. Kolejna rzecz to kwestia dotycząca tego, o czym pani minister mówiła, czyli ochrony, szczególnie turystyki, branży turystycznej. A my mamy takie pytanie: Co z firmami transportowymi?

I ostatnia kwestia: Czy rząd w jakikolwiek sposób planuje rekompensatę dla samorządów wynikającą z obniżenia podatków PIT i CIT, czyli wynikającą z mniejszych wpływów do budżetów samorządowych? Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie marszałku. Panie Premierze! Pierwsze pytanie do pana oraz do pani minister Emilewicz: Czy znają państwo treść rozporządzeń, które wydał minister zdrowia, o ogłoszeniu stanu epidemii, najpierw zagrożenia, a potem stanu epidemii, 13 i 20 marca?

Dlaczego więc dla tych firm nie ma rozwiązań o umorzeniu ZUS-u i umorzeniu podatków, skoro ich działalność została ograniczona i ich kłopoty finansowe są skutkiem decyzji, decyzji zasadnej, ale rządowej? Drugie pytanie. Wierzy pan w to. Ale jeżeli się tylko prolonguje dzisiaj daniny publiczne, składki ZUS, podatki od nieruchomości, CIT, PIT, jeżeli kredyt jest prolongowany, wielka umowa pomiędzy związkiem banków a panem prezydentem o prolongacie, a nie o odstąpieniu od rat kredytu, i skumuluje się to za kilka miesięcy, jeżeli chodzi o konieczność zapłacenia, to nie będzie żadnego odbicia ani w formie „U”, ani w postaci „V”, tylko będzie ruina w przypadku polskich przedsiębiorstw. I ostatnie pytanie, panie premierze. Unia Europejska. Czy słyszał pan o tym, że wczoraj Parlament Europejski przyjął pakiet, a więc wcześniej niż my przyjmujemy?

Otóż wczoraj wpłynął projekt ustawy, kilkadziesiąt stron, a dzisiaj do niego wpłynęła już autopoprawka, też dużo stron. To nie jest żadna tarcza, panie premierze, to jest po prostu sito, które będziemy łatać wielokrotnie. Będziemy się jeszcze nieraz spotykać, żeby kolejnym branżom pomagać. Uważam, że w takim czasie, kiedy po pandemii przychodzi tsunami w gospodarce, trzeba bardzo mocno pomagać przedsiębiorcom, nie tylko tym najmniejszym, ale tym, którzy zatrudniają większą liczbę ludzi. Tym ludziom, tym firmom nie chcecie pomóc. Wielu z nich dzisiaj i w poniedziałek podejmie decyzję, że zwolni pracowników, bo niestety w tych projektach nie ma dla nich pomocy, i to jest bardzo przykre. Tsunami w gospodarce nadejdzie w najbliższych tygodniach, ponieważ miliony ludzi mogą stracić pracę, bo wy nie chcecie im pomóc. Pomagacie bankom, chcecie pomoc kierować przez banki, a nie do firm. Dlaczego nie chcecie pomóc ratownikom medycznym, pielęgniarkom, tym, którzy pracują na pierwszej linii frontu? Wszyscy ci, którzy dzisiaj narażają życie, żeby coraz mniej ludzi było zakażonych, powinni wiedzieć, że polskie państwo o nich nie zapomni, a wy chcecie im dać przymus pracy, a nie pomoc finansową. I to jest przykre, że tak dzisiaj zachowuje się nasza wspólnota.

Panie Premierze! Wysoka Izbo! Jestem, panie premierze, szczególnie zasmucony, a właściwie chyba zażenowany tym, że polski premier powtarza przekaz rosyjskiej propagandy, że Unia Europejska nie pomaga. To jest wyjątkowo niebezpieczne, szczególnie że jesteśmy członkiem Wspólnoty. Pan, panie premierze, ma za sobą ma dwie flagi: flagę Rzeczypospolitej Polskiej, ale również flagę Unii Europejskiej. Chciałbym wiedzieć, dlaczego pan kłamie. To pieniądze, które by przepadły. Dlaczego pan kłamie, panie premierze, w taki dzień, kiedy wszyscy powinniśmy być razem? To są pieniądze, które już polski rząd może wydawać. Mówi pan, że Unia nie pomaga, tak? Moment, sprawdźmy. Uwaga, Polska nie skorzystała z unijnego mechanizmu, żeby Polacy mogli wrócić do domów za darmo. Ludzie płacili tysiące złotych LOT-owi, żeby mogli wrócić do Polski, bo Polska nie skorzystała z unijnego mechanizmu, w przypadku którego ludzie mogli wrócić do domów za darmo. Unia nie pomaga, tak? To sprawdźmy. Już otwarto oferty w tej sprawie. Ale Polska nie wzięła udziału w tym mechanizmie, bo zgłosiła się do tego przetargu zbyt późno. To jest dzisiaj problem.

Panie i Panowie Posłowie!

I muszę powiedzieć, że jestem wstrząśnięta zakresem pomocy publicznej, jakiej chciałyby udzielić kluby opozycyjne.

Chciałabym przypomnieć cytaty z państwa wystąpień, kiedy nasz rząd proponował programy społeczne takie jak 500+ oraz następnie rozszerzenie tego programu na pierwsze dziecko.

Kontrolę tę będą prowadzili - w porozumieniu - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, minister właściwy do spraw gospodarki oraz minister zdrowia. Decyzje w zależności od produktów będą podejmowane przez właściwe organy i służby.

Dziękujemy także za uwagi dotyczące możliwości korzystania z zasiłku przez osoby objęte ubezpieczeniem rolniczym, te, które są na kwarantannie, czy też możliwości rozszerzenia zasiłku opiekuńczego właśnie na tych, którzy są objęci tym ubezpieczeniem. Pani poseł Janyska w swoim retorycznym wystąpieniu pyta, czy tarcza nie starcza.

Nie chciałabym się porównywać z takimi państwami jak Dania, do której państwo się odnosili, choć nawet tam nie jest gwarantowane minimalne wynagrodzenie - mówimy o wynagrodzeniu na poziomie 75%. Nie mówimy o państwach, które miały okazję budować bogactwo swoich narodów przez minione dwa stulecia. My odbudowujemy je z mozołem przez ostatnie trzy dekady i rzeczywiście dzisiaj być może nie jesteśmy w stanie zaoferować tak szerokich programów. Bardzo często mówili państwo: zróbcie nam w Warszawie Budapeszt, a my robimy w Warszawie Warszawę w znacznie większej skali. Proszę przeczytać z uwagą rozporządzenia węgierskie, jaka tam jest proponowana dziś pomoc publiczna. Jest, owszem, zniesienie składek na ubezpieczenia społeczne. Powszechne? Nie, dla wybranych sześciu branż. Jest odroczenie, nie anulacja - odroczenie składek na ubezpieczenia społeczne. My proponujemy znacznie więcej niż inne pakiety osłonowe, które są proponowane nie tylko w państwach naszego regionu, ale także w Unii, w innych państwach członkowskich.

Ci, którzy pracują na umowach zlecenia, ci, którzy pracują na umowach o dzieło, w naszym pakiecie będą mogli uzyskać świadczenia. Oczywiście łatwo jest mówić o tym, że dziś państwo powinno wypłacić wszystkie pensje. Jak zestawić te państwa wypowiedzi z tymi w czasie minionej kadencji, kiedy mówili państwo do nas, że nie rozumiemy wolnego rynku, że wprowadzamy gospodarkę centralnie planowaną?

Pan poseł Wieczorek pyta, czy analizujemy sytuację na rynku pracy. Monitorujemy wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, ale także kontaktując się bezpośrednio z branżą, jak wygląda dzisiaj obecność pracowników na rynku pracy, z jakich świadczeń i zasiłków korzystają.

Czy planujemy rekompensaty dla samorządów? Szanowni państwo, ta ustawa jest bardzo duża, ona ingeruje w wiele elementów - oferuje nie tylko pomoc bezpośrednią, ale także ułatwienia administracyjne. Ale już w tym tygodniu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wspólnie z Ministerstwem Finansów przygotowało... analizuje, spotyka się ze Związkiem Miast Polskich, związkiem metropolii i przygotowuje, także wspólnie z samorządem, pakiet ochronny, bo zdajemy sobie sprawę, jak istotne i trudne są w tej chwili momenty, także dla samorządu. Mogą państwo powiedzieć: Czy ten pakiet wystarcza? Ja powiem tak: pewnie nikt dzisiaj nie jest w stanie powiedzieć, jaki pakiet byłby wystarczający. Musimy obserwować sytuację i reagować adekwatnie, i jesteśmy gotowi na takie działania.

Ale nie chce. Dziękuję bardzo.

Do głosowania nad tymi wnioskami przystąpimy za chwilę.

Jednak pewne rzeczy musimy sobie powiedzieć, pani minister, i dlatego musimy złożyć sprzeciw wobec wniosku PiS, żeby przejść dalej bez dyskusji, bo nic nie wiemy o podstawowych kwestiach.

Jak można debatować o skutkach ekonomicznych, kiedy pani nie podaje podstawowych informacji? Proszę państwa, w związku z tym, że został zgłoszony wniosek formalny. Czy mam tak rozumieć?

Panie pośle, 10 minut.

Bardzo proszę, po tej przerwie przystąpimy do głosowania, ponieważ zgłoszono wniosek formalny, żeby nie przystępować od razu do drugiego czytania. Za 10 minut będziemy głosować

Wznawiam obrady. W dyskusji zgłoszono wnioski o przystąpienie niezwłocznie do drugiego czytania projektów ustaw zawartych w drukach nr 299, 299-A, 301, 301-A i 302 i o skierowanie tych projektów ustaw do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Zdrowia. Pod głosowanie poddam propozycję niezwłocznego przystąpienia do drugiego czytania projektów ustaw. Jej odrzucenie spowoduje skierowanie tych projektów ustaw do komisji. I jeszcze jedna uwaga do państwa posłów na sali plenarnej. Informuję panie i panów posłów obecnych na sali plenarnej, iż w przypadku, gdy ktoś z państwa zagłosuje zarówno przy użyciu systemu do głosowania na sali, jak i przy pomocy tabletu w głosowaniu zdalnym, ważnym głosem jest głos oddany w systemie głosowania na sali, więc jeżeli ktoś próbuje głosować i.

Bardzo proszę o jej wysłuchanie. Pod głosowanie poddam zatem propozycję niezwłocznego przystąpienia do drugiego czytania wszystkich trzech projektów ustaw. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za propozycją niezwłocznego przystąpienia do drugiego czytania projektów ustaw zawartych w drukach nr 299, 299-A, 301, 301-A i 302, zechce nacisnąć przycisk.

Mogę państwa posłów prosić o to, żeby takie uwagi zostawić dla

przeciw, 2 się wstrzymało. Sejm przyjął wniosek, a tym samym wyraził zgodę na przystąpienie niezwłocznie do drugiego czytania tych projektów ustaw. Przystępujemy do drugiego czytania projektów ustaw. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie zabrać głos w drugim czytaniu tych projektów ustaw? Bardzo proszę, pan poseł Borys Budka, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Ekspresowe tempo prac. Nie ma czasu na omówienie wszystkich poprawek, które będziemy zgłaszać. Tak jak obiecaliśmy, przez ostatnie tygodnie konsultowaliśmy to z wami, przedsiębiorcami, pracownikami, ludźmi służby zdrowia, z wami, którzy na co dzień pomagacie Polakom i którzy na co dzień borykacie się z problemami koronawirusa, borykacie się również z wielkim strachem o waszą przyszłość, o przyszłość waszych rodzin. Dlatego składamy kilkadziesiąt poprawek, które sprawią, że ta dziurawa, tekturowa tarcza antykryzysowa może stać się rzeczywiście (Dzwonek) narzędziem, które będzie was chronić. Szanowny Panie Premierze! To jest test dla pana. to jest test na pana wiarygodność. Jeden test oblewa pan od dłuższego czasu. Nie wprowadzając stanu nadzwyczajnego, nie daje pan możliwości ubiegania się o odszkodowania tym setkom tysięcy ludzi, [[Oklaski]] którzy na co dzień dotknięci są właśnie waszymi decyzjami. W naszych poprawkach gwarantujemy rezygnację ze składek ZUS bez wyjątku dla wszystkich przedsiębiorców, którzy są dotknięci koronawirusem, skutkami tej epidemii, ale również dla pracowników wszystkich branż bez względu na to, jaka jest wielkość pracodawcy, jaka jest skala działalności gospodarczej i rodzaj tej działalności. Gwarantujemy minimalne wynagrodzenia z budżetu państwa. Mówiliście o braku deficytu. Oświadczenie przedsiębiorcy ma być podstawą do udzielenia pomocy. Dzisiaj zajmujecie kolejne rachunki bankowe, dzisiaj prowadzicie kolejne egzekucje administracyjne. Czas najwyższy powiedzieć: stop. Oświadczenie przedsiębiorcy ma być podstawą do udzielenia tej pomocy. Szybki, 3-dniowy zwrot podatku VAT. Pracodawcy potrzebują tych pieniędzy, by wypłacać wynagrodzenia. Wy je przetrzymujecie na rachunkach Skarbu Państwa. 20 mld na służbę zdrowia. Konkrety. Z pieniędzy europejskich przeznaczmy to właśnie dla tych, którzy na co dzień walczą z koronawirusem, na środki ochrony osobistej, na wyposażenie szpitali. 2 mld daliście na TVP, 20 mld chcemy dać na służę zdrowia. Zasiłek opiekuńczy dla was, drodzy rodzice, którzy od poniedziałku znowu będziecie ze swoimi pociechami, dlatego że nie będą chodziły do szkół, przedszkoli i żłobków, ale również dla tych, których dzieci mają powyżej 8 lat. Co macie zrobić? Co macie zrobić, jeśli wasze dzieci nie mają opieki? Co macie zrobić, jeśli zostaniecie bez środków do życia? Gwarantujemy naszą poprawką pomoc dla was. Elastyczny czas pracy to podstawa, by szybko reagować na zmieniające się warunki. Obniżenie czynszów dla lokali zarówno gastronomicznych, jak i handlowych, bo tam po prostu nie może być prowadzona działalność gospodarcza. Gwarancje bankowe dla wszystkich firm bez wyjątku, bez dzielenia na branże, bez kategorii lepszego i gorszego sortu. Bardzo istotne jest to, żeby móc reagować bardzo szybko. Te kilkadziesiąt poprawek chcielibyśmy omówić szczegółowo, chcielibyśmy pokazać, jakie konkretne rozwiązania są przez nas przedstawianie, ale niestety wprowadzono taki tryb pracy, szanowni państwo. Dzisiaj jesteście albo w waszych domach, albo w waszych miejscach pracy i oczekujecie rzetelnej pracy od nas, parlamentarzystów. Tymczasem nie ma pracy w komisjach, nie ma merytorycznej pracy nad tym, co zgłaszamy. To jest kilkadziesiąt stron dobrych poprawek. Dziękuję wam wszystkim, którzy zgłaszaliście te postulaty. Dziękuję zarówno pani ze sklepu spożywczego, która powiedziała, że przychód nie może być kategorią, która będzie różnicować przedsiębiorców, bo ona przychód ma duży, ale będzie miała stratę. Dziękuję związkom pracodawców. Dziękuję wam, zwykłym ludziom, którzy boicie się o waszą przyszłość. Wasze poprawki uwzględniliśmy, bo wy jesteście dzisiaj najważniejsi. I raz jeszcze podkreślam: to jest test na solidarność społeczną, ale to jest również test na to, czy wreszcie będziemy wspólnotą, czy wreszcie rząd przestanie dzielić na lepszy i gorszy sort. Dziś mówimy: sprawdzam. Dziś, panie premierze, mówimy: sprawdzam, ale, kochani, pana premiera nie ma, pan premier wyszedł. I właśnie tak wygląda ten dialog, wspólnota, to, o czym zapewniał rząd. Szanowni Państwo!

Bardzo proszę, pan poseł Maciej Konieczny, klub parlamentarny Lewica. Proszę państwa, czas był prawie dwukrotnie przekroczony, więc.

Wysoka Izbo! Codziennie docierają do nas setki wiadomości od polskich pracowników o tym, jak łamane są ich prawa, jak narażane jest ich zdrowie, jak z dnia na dzień ludzie tracą środki do życia. Jedna historia powtarza się często. W obliczu zagrożenia wirusem szef stawia przed bramą zakładu człowieka z termometrem i ten człowiek mierzy temperaturę: raz na czole, raz na nosie, raz na ręce, raz na kurtce. Jak jest za dużo ludzi, to nie mierzy w ogóle. Dlaczego o tym mówię? Dlatego że tarcza antykryzysowa, te działania rządu przypominają mi tego człowieka z termometrem. Zamiast realnie pomóc, rząd udaje, że coś robi. Panie Premierze! To nie jest czas na udawanie. Nadchodzi kryzys gospodarczy, jakiego świat nie widział. Znaczna część naszej gospodarki, znaczna część światowej gospodarki musi stanąć, bo od tego zależy zdrowie i życie naszych bliskich. Albo państwo stanie na wysokości zadania i będą odważne działania, albo z tego kryzysu łatwo się nie wygrzebiemy. Rządowi odwagi zabrakło. Zamiast pomóc pracownikom, bezrobotnym, drobnym przedsiębiorcom, Mateusz Morawiecki proponuje radykalne cięcia płac, wydłużenie czasu pracy i bardzo skromne zapomogi. To gospodarcze samobójstwo. Polacy muszą mieć pieniądze w kieszeni, żeby kupować towary i usługi. Polacy nie mogą zostać jedynie z długami, bo wtedy z tej recesji nie wyjdziemy przez lata. Te rozwiązania proponowane przez rząd tylko nakręcą spiralę recesji. Tarcza antykryzysowa nie chroni pracowników i wbrew temu, co mówiła minister Emilewicz, tego samego zdania są związki zawodowe. Dziś miliony osób na śmieciówkach z dnia na dzień tracą środki do życia. Zamiast realnego wsparcia dostają jednorazową zapomogę. To kpina. Każdy pracownik i każda pracownica, bez względu na charakter umowy, muszą mieć zagwarantowany dochód, minimum płacę minimalną albo więcej. Tego domaga się Lewica. Wraz z kryzysem wróci wysokie bezrobocie. Tymczasem polski system wsparcia dla bezrobotnych to od dawna jest kpina. Bardzo skromne, niewystarczające zasiłki, które do tego trafiają jedynie do garstki osób. A co rząd proponuje bezrobotnym, tym obecnym i przyszłym? Nie zaklinajcie rzeczywistości. Bezrobocie na wielką skalę już puka do naszych drzwi. Wybór jest prosty: albo prawdziwy system wsparcia dla bezrobotnych, albo tymczasowy dochód gwarantowany dla wszystkich. To nie jest czas na tchórzliwe półśrodki. Rząd musi wesprzeć polskie przedsiębiorstwa - to jest oczywiste - tak żeby chronić polskie miejsca pracy, ale ta pomoc musi być prawdziwa. Te rozwiązania, które zaproponowaliście, nie uratują miejsc pracy w Polsce. Wzorem Danii Lewica proponuje 75% dopłaty od państwa, ale pod dwoma warunkami: żadnych zwolnień i żadnych obniżek wynagrodzeń. Położyliśmy konkretne, duńskie rozwiązania na stole. Usłyszeliśmy od minister Emilewicz, że ich nie wprowadzi. Pani Minister! Polski nie stać na masowe bankructwa polskich przedsiębiorstw. Polski nie stać na masowe bezrobocie. Polski nie stać przede wszystkim na radykalny spadek dochodów Polaków. Usłyszeliśmy, że rząd nie ma na to pieniędzy, ale 70 mld dla banków pani minister jakoś znalazła. Dla bezrobotnych pieniędzy nie ma, dla pracowników pieniędzy nie ma, ale dla banków są. Co zrobiły banki? Skróciły czas spłaty kredytu, tak że raty są większe, a banki jeszcze na tym zarobią. W ogóle co to jest za sytuacja? Prezydent Rzeczypospolitej prosi banki o łaskę. Kto tu tak naprawdę rządzi? Banki są dla pana premiera, dla obecnego rządu dziesięć razy ważniejsze niż pracownicy ochrony zdrowia. Banki są ważniejsze niż ci, którzy dzisiaj realnie walczą z koronawirusem. Dla lekarzy, dla pielęgniarek w tych ustawach jest tylko przymus i więcej pracy. Całe szczęście, że dzięki Lewicy udało się z tej ustawy usunąć najbardziej skandaliczny zapis, taki, żeby państwo mogło zmuszać lekarzy do pracy właściwie bez końca. Personel medyczny naprawdę nie potrzebuje więcej podziękowań, nie potrzebuje żadnych specjalnych uchwał, w których Sejm oddaje im cześć. Personel medyczny potrzebuje godnych płac, godnych warunków pracy (Dzwonek) i ochrony zdrowia, która działa. Tę tarczę można jeszcze uratować. Składamy dziesiątki poprawek, które zabezpieczą pracowników, bezrobotnych, małe firmy, pomogą lekarzom i pielęgniarkom. Wyciągamy rękę i kładziemy na stole konkretne rozwiązania, ale chcemy powiedzieć jasno: jeżeli te poprawki nie zostaną przyjęte, koalicyjny klub Lewicy zagłosuje przeciw. Dziękuję, panie pośle. Proszę bardzo, pan poseł Władysław Kosiniak-Kamysz, Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15. Wysoka Izbo! Część już zgłaszaliśmy w pierwszym czytaniu. Zacznę od spraw najważniejszych. Po pierwsze, życie i zdrowie, bo nie ma sprawy ważniejszej niż ochrona życia, ochrona zdrowia, wsparcie dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia. Dziękuję za te poprawki, które już były omawiane, dotyczące lepszego wynagrodzenia pracowników, tych, którzy dzisiaj są na pierwszej linii walki.

Dzisiaj jest wiele firm odzieżowych, które wyhamowały produkcję, bo nie mają rynku zbytu. One są gotowe podjąć i przestawić swoją produkcję na sprzęt ochrony medycznej dla szpitali, również dla jednostek pomocy społecznej czy służb mundurowych, tylko trzeba do tego włączyć Agencję Rezerw Materiałowych, żeby dała gwarancję i zabezpieczyła odebranie tego wszystkiego, co będą wytwarzać polskie firmy odzieżowe, nie tylko odzieżowe, ale też produkujące różnego rodzaju sprzęt, który może być dzisiaj wykorzystywany do ochrony. Dobrze, że jest transport z Chin, ale powinno być tu zabezpieczenie. Kolejna sprawa. Bez płynności nie uratujemy polskich firm. Chodzi o złożoną przez marszałka Tyszkę propozycję dotyczącą funduszu płynności, funduszu, który będzie otwartą linią kredytową o gigantycznych rozmiarach, bo takie muszą być. To nie mogą być pożyczki 5 tys. z Funduszu Pracy.

Firmy, które stracą płynność finansową, zaraz upadną, zwolnią wszystkich pracowników. Wtedy już im nawet najlepsze świadczenia socjalne nie pomogą, bo one nie zastąpią miejsca pracy. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że dzisiaj inwestycja dla firmy to jest inwestycja dla prowadzącego działalność gospodarczą, ale również dla pracownika. Szkoda, że nie prowadziliście autentycznego dialogu ze związkami i z pracodawcami w ramach Rady Dialogu Społecznego.

Kolejne kwestie, bardzo merytoryczne, dotyczące - jeszcze raz powtórzę - dobrowolnego ZUS-u, zwolnienia z CIT-u, z PIT-u. Jeżeli tego nie zrobimy, to w październiku, w listopadzie tych firm po prostu nie będzie i o żadne daniny publiczne już nie będziemy mogli wnioskować. Upominam się po raz kolejny o rolników. Na posiedzeniu Rady Gabinetowej w pierwszej wersji pakietu antykryzysowego - to też dla jasności dla tych, co nas oglądają - nie było, moi drodzy, ani słowa o rolnikach, o gospodarstwach rolnych, o przemyśle rolno-spożywczym. Liczę, że rolnicy objęci kwarantanną będą mieli prawo do minimalnego wynagrodzenia. Bardzo ważne jest wsparcie polskiego rzemiosła. To są firmy, to są tradycyjne warsztaty, które utrzymywały polską gospodarkę zawsze, w najtrudniejszych czasach.

W ten sposób poszerzymy krąg osób, które są uprawnione do zapłacenia przez państwo ZUS-u za nich, i więcej firm z tego skorzysta. Dziękujemy za wszystkie wnioski. Przedstawiamy je w naszych poprawkach. Dotyczą one i świadczeń socjalnych, i dodatkowego zasiłku dla osób opiekujących się dziećmi, dodatkowego wsparcia dla tych wszystkich, którzy idą do pracy, a ktoś musi zostać w domu i rodzice muszą się dzielić tymi obowiązkami. Tu nie może być granicy 8 lat, bo czym się różni opieka nad ośmiolatkiem czy dziewięciolatkiem. 12 lat, 15 lat - to są te granice, które powinny być. Wysoka Izbo! Solidarność jest zasadą dwukierunkową. Tylko wtedy jesteśmy w stanie uratować polską gospodarkę. Tu jest cały pakiet rozwiązań dla samorządów. Jeżeli rząd nie będzie rekompensował im czynszu, który umorzy, podatku od nieruchomości, który umorzy, czy podatku rolnego, wspólnoty samorządowe tego nie wytrzymają. Staną wszystkie inwestycje. Trzeba się też zastanowić nad kolejnymi ruchami w następnych latach. Czy dzisiaj jest nam potrzebny Centralny Port Komunikacyjny?

Bez miejsc pracy, bez naszego bezpieczeństwa tak naprawdę wszystko inne zejdzie na dalszy plan. Liczymy, ze ta ustawa będzie wielokrotnie modyfikowana. Szczególnie liczymy na otwartą, wysoką linię kredytową, fundusz płynności w Banku Gospodarstwa Krajowego. On musi powstać.

Pani Marszałek!

Zastanawiam się, dlaczego co miesiąc nie ma jakiejś epidemii. Moglibyśmy uchwalać wspaniałe ustawy, które pomogą przemysłowi, ludziom pracy. Dlaczego tego nie robimy? Zwykły, szary człowiek, zapłaci 38 mln konsumentów, bo lewica dba o ludzi pracy, a prawica dba o konsumentów.

A na zakończenie, Wysoka Izbo, postanowiłem, dopóki koronawirus nie opuści polskich ziem, się nie golić. Mam nadzieje, że nie położą mnie do grobu z długą, siwą brodą, która by mi muszkę zakryła. Dziękuję, panie pośle.

Ile zostało czasu? Wysoka Izbo!

Dlaczego w projekcie jest założenie, że będziemy wspierać także te zagraniczne wielkie korporacje, które mają swoje siedziby nie tylko poza Unią Europejska, przepraszam, nie tylko poza Polską, ale także poza Unią Europejską? Niech te korporacje zgłaszają się do swoich rządów. My zadbajmy dzisiaj o polskiego przedsiębiorcę i tym samym o polskiego pracownika. Pamiętajmy też, że jest kolejny haczyk w tej nowej ustawie, czyli przedłużenie, automatyczne przedłużenie pozwoleń o pracę dla cudzoziemców. Co będzie, jak już gospodarka naprawdę stanie i Polacy zaczną tracić pracę, a cudzoziemcy dalej będą mogli tutaj pracować? Kto będzie miał największy problem? Nasi obywatele. Zadbajmy o nich w pierwszej kolejności. Dlatego koło Konfederacja zgłasza do wszystkich trzech projektów swoje poprawki. Dziękuję. Bardzo proszę. To się nie uda, to się musi wywalić. Nie można bezkarnie uchwalać setek stron przepisów w takich warunkach, w takim pośpiechu. Do walki z epidemią trzeba być dobrze przygotowanym, trzeba mieć przemyślane ustawy i procedury, a wy robicie jakąś wielką improwizację, wykonujecie setki chaotycznych ruchów bez ładu i składu. My też tak poprawiamy jeden bubel prawny kolejnym bublem prawnym, bo nie mamy czasu tego spokojnie przemyśleć.

Opozycja, która te specustawę poprzednio lekkomyślnie przyklepała zwiedziona kilkoma poprawkami przyjętymi na swoją korzyść, dopiero po 2 tygodniach się zorientowała, że głównym powodem uchwalenia tej ustawy było tak naprawdę wprowadzenie stanu wyjątkowego bez odkładania wyborów. Nie wolno przyklepywać i żyrować w ciemno jakiejś prowizorki tworzonej przez rząd na kolanie. Powiedziałem, że skutek będzie taki, że po prostu zabraknie maseczek. Oczywiście tak się stało.

Więc co najlepszego zrobiliście, kto miał wtedy rację? Oczekuję w tym momencie na oklaski. Chyba się należą za udane proroctwo, prawda? Kiedy dramatycznie brakuje maseczek, szykujecie jakiś tam geszeft, po prostu próbując zagwarantować monopol zaprzyjaźnionej firmie i interweniując w zagranicznych serwisach, żeby przyblokowały prywatne zakupy Polaków. Czego się z tego nauczyliście?

Wszelkie regulacje, wszelkie reglamentacje, regulowane ceny to jest zaproszenie biedy do stołu. Czego się nauczyliście? Lista posłów zapisanych do głosu została. Bardzo proszę.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Otóż jest niewątpliwym - nie chcę użyć słowa: kłamstwem - wynikiem braku, jak rozumiem, umiejętności czytania aktów prawnych stwierdzenie, jakoby te ustawy miały gwarantować raptem kilka mld zł ze strony czy to budżetu, czy to w ogóle sektora finansów publicznych, bo na to spójrzmy.

To z samego sektora finansów publicznych.

Tak że miejmy tego świadomość i bardzo proszę o niewprowadzanie opinii publicznej w błąd.

Powiem o najważniejszych z nich. Najważniejsza sprawa z tego pakietu to jest kwestia związana z tym, żeby dla samozatrudnionych, dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Myślę, że jeśli chodzi o niektóre rzeczy, będę także rekomendował mojemu klubowi poparcie niektórych poprawek opozycji, bo pojawiają się także i dobre pomysły. Z niezrozumiałych powodów część przedstawicieli opozycji bardzo się zdenerwowała jakąś metaforą użytą w moim wystąpieniu podczas pierwszego czytania. Pan przewodniczący Kosiniak aż się zatrząsł.

Dziękuję bardzo. Dobrze, sprostowanie. Bardzo proszę, pan poseł Władysław Kosiniak-Kamysz.

Ma pan zadanie jako minister, szef komitetu stałego, to proszę je wykonywać. A o historii z chęcią podyskutujemy, tylko to nie jest ten czas.

Dziękuję, panie pośle. O głos poprosiła pani minister Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju. Bardzo proszę.

Tak jak mówiliśmy na początku, nie ma dzisiaj osoby, nie ma dzisiaj organu, nie ma dzisiaj podmiotu, nie ma przedsiębiorstwa, które nie muszą mierzyć się z tymi konsekwencjami. W tych rozwiązaniach, które przygotowaliśmy, dotknęliśmy - odrobinę - kwestii związanych z prawidłowością funkcjonowania samorządu, z tym, aby samorządy nie zostały sparaliżowane w związku z ograniczeniami.

Tak jak wspominałam wcześniej, my proponujemy inne rozwiązania - na miarę naszych możliwości i na miarę potrzeb i sytuacji, w której się dzisiaj znajdujemy. Ale dzisiaj apelujemy do państwa: przyjmijmy te rozwiązania, bo one są potrzebne przedsiębiorcom i pracownikom jak najszybciej, po to aby w ten 1 kwietnia mogli wejść z pewnością utrzymanych miejsc pracy. Panie pośle, proszę mi powiedzieć, którzy ekonomiści na świecie są przygotowani do kryzysów, które mają nadejść. Zawsze jesteśmy świetnie przygotowani do tych, które się zakończyły. Ta ustawa nie jest arcydziełem legislacyjnym, to prawda. I w tym pośpiechu, w tym zbieraniu wielu spraw, które trafiały do nas od przedsiębiorców, pewnie nie napisaliśmy doskonałej legislacyjnie ustawy, ale jestem przekonana, że przygotowaliśmy dobre przepisy, które uratują miejsca pracy, które uratują polskie firmy. Tak, popełniamy być może czasami błędy i jesteśmy gotowi się do nich przyznać. Tak, dziękowaliśmy tym, którzy zwrócili nam uwagę na to, że formularz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ma 11 stron, potem 4 strony, kiedy prosimy o odroczenie składek na ubezpieczenia społeczne. Wymagało to kontaktu z Komisją Europejską, zmiany schematu pomocy de minimis i następnie krótkiej pracy informatycznej - w ciągu jednego weekendu. Od poniedziałku ten formularz ma niespełna 1 stronę, jest naprawdę prostym oświadczeniem. Taka jest nasza ustawa. Chciałabym, żebyśmy na tej wojnie stanęli ramię w ramię, a nie przeciwko sobie. Walczmy z wirusem, a nie walczmy ze sobą nawzajem. Zamykam dyskusję. Nie, panie pośle. Zamykam dyskusję. Nie, panie pośle, to nie było odwołanie się tylko do pana, tylko do wszystkich państwa, którzy zabierali głos.

W związku z tym, że w drugim czytaniu zgłoszono do projektu ustawy poprawki - tych poprawek jest, proszę państwa, 257 - proponuję, aby Sejm przystąpił do trzeciego czytania projektu ustawy po doręczeniu paniom i panom posłom zestawienia poprawek. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę.

Będziecie państwo wtedy informowani SMS-ami.